Nie chcielibyśmy tego.

Może część KRS-u powinna być w wyborach powszechnych wybierana przez obywateli?

Opowiadamy się za jej odrzuceniem. Pan poseł Krystian Kamiński, koło Konfederacji.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kto miał czas zapoznać się z poprawkami w tak ważnej ustawie? Dobrze wiemy, że nikt, ale dla państwa z PiS naturalnie to nie ma znaczenia. Proponowane zmiany ustawy to tylko i wyłącznie następna odsłona walki o wpływy między partią rządzącą a władzą sądowniczą. Wbrew temu, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, nie ma dziś łatwego rozwiązania tej sytuacji. Jednak również wbrew temu, co mówi totalna opozycja, nie ma dziś zgody na dalsze trwanie w tak niewydolnym systemie sądowniczym, w którym zwykli obywatele nie mają poczucia sprawiedliwości, a przedsiębiorcy na wyrok muszą czekać latami. Wszyscy widzimy, że potrzebna jest dziś gruntowna reforma systemowa, tak aby usprawnić nasze sądy, aby uczynić je przyjaznymi dla obywateli. Sądy powinny być przede wszystkim szybkie i sprawiedliwe. Sędziów trzeba uwolnić od wykonywania niemerytorycznych, biurokratycznych zadań. Właśnie dlatego jako Konfederacja proponujemy parametryzację sądów, przypisywanie asystentów na stałe do każdego sędziego, elektroniczny obieg dokumentów, a docelowo - proces w 1 miesiąc. To są reformy, na które czekają Polacy. Aby jednak rozwiązać obecny kryzys sądownictwa, którego jesteśmy świadkami, potrzebujemy rozwiązań systemowych. Dlatego Konfederacja również zaproponuje zmiany ustrojowe przecinające konflikty personalne. Musimy wszyscy zrobić krok w tył i rozpocząć debatę nad resetem konstytucyjnym, nad zmianą konstytucyjną, która rozwiąże ten chaos spowodowany zarówno przez Platformę Obywatelską, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość. Warto też zastanowić się nad możliwością dopuszczenia w szczególnych przypadkach ławy przysięgłych, aby surowość wyroku odzwierciedlała poczucie społecznej krzywdy. Naszym zdaniem pora rozpocząć szeroką debatę nad polskim sądownictwem. Inaczej takie przepychanki, których jesteśmy świadkami, będą nam towarzyszyć jeszcze bardzo długo. Teraz głos ma pan poseł Robert Winnicki, również koło Konfederacji. Wysoka Izbo! Po pierwsze, trzeba jasno powiedzieć Komisji Europejskiej: Wara od polskiego stanowienia prawa, od tego, co robi suwerenny Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Nie macie prawa wtrącać się w naszą wewnętrzną debatę. Nie macie prawa do tego, żeby z Brukseli dyktować, w jaki sposób będzie wyglądało polskie sądownictwo, polskie prawo. I to dzisiaj musi paść z tej mównicy bardzo jasno. Druga sprawa to to, jak wygląda polskie sądownictwo, jak wyglądało w 2015 r., jak wyglądało wcześniej. Niestety sytuacja tam jest po prostu zabagniona. Jest to bagno znaczącej niesprawiedliwości, ciągnących się procesów, nieskuteczności, krzywdzących wyroków. Jest i coś, o czym oczywiście mówią też niektórzy spośród sędziów - że są nadzwyczajną kastą. Nie istnieje i nie istniał wcześniej de facto realny trójpodział władzy, tak by w jakikolwiek sposób kontrolowana była władza sądownicza. Problem polega na tym, że do tego bagna, zamiast go osuszać przez 4 lata, zamiast osuszać bagno polskiego systemu sądowniczego przez 4 lata, wyście wpuścili swoją rurę i sądzicie, że jak dolejecie trochę od siebie, to bagno to wyschnie. Otóż nie, nie wyschnie, śmierdzi jeszcze bardziej. I z tą właśnie sytuacją dzisiaj się zderzamy, mierzymy. Ta łata, o której mówił pan poseł Czarnek. Robicie łatę na łacie, 4 lata łatania i jakby sytuacja, ten materiał, który łatacie, nie wygląda lepiej. Wygląda to coraz gorzej, coraz mniej sprawnie. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty. Podeszliście do tematu nie od strony reform systemowych, strukturalnych, tylko kadrowych.

W złym systemie wpuszczenie tam nawet znacznej liczby osób, których zresztą nie macie za dużo, tych kadr, żeby ten system sądowniczy uzdrowić, nie powoduje jego uzdrowienia. Taka jest sytuacja. I możecie tych reform jeszcze namnożyć 500 i może trwać to jeszcze dekady i systemu nie uzdrowicie. Jesteście totalnie nieudolni, niekompetentni i dlatego Konfederacja nie będzie popierała tego projektu ustawy.

Teraz przystępujemy do kolejnych elementów tej debaty.

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Szanowne Panie Posłanki i Szanowni Panowie Posłowie! Jako rzecznik praw obywatelskich mam obowiązek stać na straży praw i wolności człowieka i obywatela. Prawo do sądu, a w szczególności prawo do niezależnego sądu, to jedno z praw określonych w konstytucji w art. 45 oraz w umowach międzynarodowych, które Polska ratyfikowała. Z różnych powodów oraz za pomocą różnych środków prawnych prawo do niezależnego sądu jest w Polsce podważane co najmniej od 4 lat. W tym czasie doczekaliśmy się jako państwo licznych krytycznych uwag ze strony organów ONZ, Rady Europy, OBWE czy Unii Europejskiej. Czterokrotnie w sprawie różnych reform, które dotyczyły naszego sądownictwa, wypowiadał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ostatnio 19 listopada 2019 r. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Komisję Europejską, dotyczącego mechanizmu dyscyplinarnego w stosunku do sędziów. Jest także zawisłych kilka pytań prejudycjalnych zadanych przez polskie sądy. Zaniepokojenie sytuacją w Polsce, jeżeli chodzi o sądownictwo, wyrażają obywatele w ramach protestów na ulicach, organizacje pozarządowe, dziekani wydziałów prawa, samorządy prawnicze, i wszystkie osoby, którym na sercu leży przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W obliczu tych zagrożeń systemu prawnego moim zdaniem powinniśmy się spodziewać podjęcia działań służących naprawieniu stanu prawnego. Powinniśmy spodziewać się podjęcia inicjatyw, szczególnie legislacyjnych, które sprowadzą Polskę na drogę praworządności, przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej oraz prawa europejskiego. Powinniśmy się spodziewać działań podejmowanych w pełnej odpowiedzialności za porządek konstytucyjny. Niestety zamiast tego obserwujemy represje w stosunku do sędziów, polegające na wszczynaniu postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych, odwoływanie z delegacji sędziowskich czy wręcz zawieszanie ich w wykonywaniu obowiązków. Obserwujemy także dyskredytowanie przedstawicieli władzy sądowniczej przez przedstawicieli innych władz. No i wreszcie obserwujemy debatę nad ustawą, która moim zdaniem pogłębi stan kryzysu praworządności. Chciałbym podkreślić, że kryzys praworządności nie jest neutralny dla obywateli oraz dla gospodarki. Wszelkie zakłócenia, jeżeli chodzi o gwarancje prawa do niezależnego sądu, będą miały wpływ na respektowanie zasady wzajemnego zaufania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemów sądowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Braku możliwości rozwiązania, zażegnania aktualnego kryzysu będzie oznaczać brak możliwości uznawania orzeczeń sądów polskich przez sądy innych państw członkowskich, a także brak możliwości współpracy z polskimi sądami. To będzie wpływało na działalność naszych sądów w kontekście spraw karnych, rodzinnych oraz cywilnych, w tym także w kontekście ochrony inwestycji. Wiemy dobrze, że procedowana ustawa ma wiele wad. Jeszcze w środę przedstawiłem kompleksową opinię na jej temat. Krytyczną opinię przedstawił także Sąd Najwyższy, jak również Biuro Analiz Sejmowych. Moim zdaniem wprowadzone w nocy poprawki nie naprawiają ustawy, co więcej, wręcz pogarszają sytuację. Chciałbym podkreślić, że mam wrażenie, że niektóre z nich w ogóle nie były konsultowane nawet z zainteresowanymi podmiotami, bo trudno się tego spodziewać między godz. 22 a godz. 5 nad ranem. Ma on być powoływany przez prezydenta. Również uprawnienie prezydenta do wskazywania osoby prowadzącej posiedzenie zgromadzenia ogólnego Sądu Najwyższego czy osoby pełniącej funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mam wrażenie. Już od kilku lat niestety obserwujemy ten tryb procedowania ustaw. Najpierw pojawia się projekt poselski, który omija etap konsultacji społecznych, następnie następuje szybki tryb procedowania w ramach prac komisji, zgłaszanie poprawek w ramach tych prac, brak możliwości rzetelnej dyskusji, wielki pośpiech. Natomiast efektem jest to, że na podstawie tej ustawy, która jest procedowana, zwiększa się znacząco uprawnienia dwóch izb Sądu Najwyższego: Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To właśnie te dwie izby zostały stworzone i obsadzone w 2018 r. przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie rekomendacji wydanych przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie i to w stosunku do tych izb można mieć poważne zastrzeżenia w świetle wyroku Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada tego roku, a także wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia tego roku w sprawie pana sędziego Andrzeja Kuby. Dlaczego akurat te dwie izby są wzmacniane o nowe kompetencje? Dlaczego Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ma mieć prawo weryfikacji innych wyroków Sądu Najwyższego, które dotyczyłyby obsady sądów? Czy to ma być kolejna izba, która ma się stać superizbą oceniającą inne izby Sądu Najwyższego? Chciałbym podkreślić, że ustawa wprowadza negatywne klauzule, które nie pozwalają na weryfikowanie, czy organ jest sądem lub czy osoba jest sędzią. I projekt w ten sposób w istocie zmierza do intencjonalnego wyłączenia spod kontroli sądowej legalności powołania i działania organów sądowych, a także legalności powołania do pełnienia urzędu sędziego. Moim zdaniem jego celem jest powstrzymanie sądów przed bezpośrednim stosowaniem zarówno wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również wyroków Sądu Najwyższego, tego który już został wydany 5 grudnia, jak również tych które są zaplanowane w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i które zgodnie z zapowiedziami mają być wydane w styczniu 2020 r. Natomiast chciałbym podkreślić, że odkąd pamiętam sędziowie posiadali autonomiczną możliwość weryfikowania składów sędziowskich. Swego czasu była taka sytuacja, kiedy sędziowie byli nieprawidłowo delegowani do sądów przez wiceministrów sprawiedliwości i to podlegało weryfikacji. Były też sytuacje, kiedy orzekali nie w tych sądach, co powinni, źle była ustawiona ich właściwość. Pojawiały się problemy z czynnościami orzeczniczymi asesorów. Każdy sędzia powinien mieć taką możliwość, a ustawa de facto taką możliwość wyłączy i będzie w ten sposób krępowała obywateli w realizacji ich praw. Obywatele nawet nie będą mogli się dopominać o weryfikację składów, skoro będą wiedzieli, że z tego tytułu będzie sędziom groziła odpowiedzialność dyscyplinarna, jeśli tylko podejmą jakiekolwiek decyzje sprzeczne z intencją ustawodawcy. Dlatego, chcąc rozwiązać doraźny problem wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, de facto dewastuje się procedury sądowe. Chciałbym także zauważyć, że tego typu rozwiązanie zmierza do pominięcia standardów konstytucyjnych oraz standardów europejskich, zmierza także do pominięcia standardów wynikających z europejskiej konwekcji praw człowieka. Co więcej, tak jak wspomniałem, jest to potwierdzane przez rozszerzenie i zaostrzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, które projektodawcy proponują. W tym kontekście bardzo niebezpieczne są te postanowienia ustawy, które odnoszą się do sfery wolności słowa oraz wolności zrzeszania się sędziów. Dla mnie jest oczywiste, że sędziowie nie mogą angażować się w działalność publiczną, której nie można pogodzić z godnością urzędu sędziego. O tym mówi konstytucja. Oczywiście sędziowie nie powinni wypowiadać się na takie tematy, jak programy socjalne rządu, obronność, polityka zagraniczna, system edukacji. A jeżeli już się wypowiadają, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy trafia do nich aktualna sprawa, która tego dotyczy, i kiedy w inny sposób, niż poprzez orzeczenie, nie mogą się wypowiedzieć. Natomiast czym innym jest wypowiadanie się na temat istoty własnego zawodu oraz niezależności sądownictwa, [[Oklaski]] bo sędziowie mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek wypowiadać się na tematy dotyczące ustroju sądownictwa, niezależności sądów, niezawisłości sędziów. Po to zostali wykształceni, aby na ten temat się wypowiadać, bo rozumieją, jak działa system prawny, ale także po to, aby czasami się bronić przed próbami ograniczenia ich statusu przez przedstawicieli innych władz. To nie jest polityka, to nie jest działalność publiczna niedająca się pogodzić z godnością urzędu. To jest działalność, która służy obronie praw obywatelskich, a w szczególności prawu do niezależnego sądu wyrażonego w konstytucji. Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panowie Posłowie! W ustawie znajdziemy szereg różnych rozwiązań, które są nowe, których nawet nie sposób było przeanalizować przez te kilka godzin od godz. 5 rano. Takie rzeczy np. jak zmiany dotyczące trybu uchylania immunitetu i uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Cały czas się zastanawiam, czemu służy art. 8 ustawy, który pozwala być może na zatwierdzanie różnych sytuacji, kiedy właśnie wyroki były wydawane przez składy nie do końca odpowiadające dotychczasowym ustawom. Prawdopodobnie z biegiem czasu dowiemy się, co tak naprawdę w tej ustawie się jeszcze znajduje. Oczywiście jako rzecznik praw obywatelskich będę szerzej projekt analizował także w kontekście poprawek, które zostały zgłoszone. Natomiast już na tym etapie uważam, że projekt ustawy narusza ustawę zasadniczą, łamie podstawowe zasady porządku prawnego. Moim zdaniem uchwalenie projektu w proponowanym kształcie zakwestionuje w istocie uczestnictwo Polski w wymiarze prawnym Unii Europejskiej i w Radzie Europy. Ostatecznie podda polskie sądy i polskich sędziów politycznej kontroli organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a co najważniejsze, drastycznie obniży poziom sądowej ochrony praw jednostek. Uważam, że przyjęcie tej ustawy to droga do prawniczego polexitu - wyjścia Polski z Unii Europejskiej w zakresie respektowania podstawowych reguł dotyczących praworządności, wydrążenia naszego członkostwa z istoty, jaką jest budowanie systemu prawnego opartego na zasadzie współpracy, wzajemnego zaufania oraz respektowania podobnych standardów dotyczących praworządności. Dziękuję.

Teraz głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan Marcin Warchoł.

Panie Rzeczniku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

W przypadku kradzieży wiertarki również półtora roku. Przez 7 miesięcy sędzia od wiertarki orzekał, wydał kilkanaście orzeczeń. Pani znowu krzyczy. To jest ta różnica pracy, jakości Izby Dyscyplinarnej w stosunku do tego, co było przed reformą. Tego się boicie? Boicie się sprawnych, szybkich wyroków. Boicie się orzekania w 1 dzień o wyrzuceniu sędziego z urzędu. Izba kontroli nadzwyczajnej, druga z izb, która została dzisiaj tutaj przez pana rzecznika wspomniana, uchyla niesprawiedliwe wyroki. Pani, która padła ofiarą lichwiarzy, po wzięciu pożyczki wysokości 15 tys., musiała oddać przeszło milion po jednym roku, 730% to koszty pozaodsetkowe. Dzięki prokuratorowi generalnemu właśnie nowo powołana izba uchyliła ten niesprawiedliwy wyrok. Panie rzeczniku, ale ile pan wniósł skarg nadzwyczajnych do izby kontroli nadzwyczajnej, jakie są pańskie sukcesy? Może pan powie wszystkim naszym obywatelom, jak pan bronił praw obywatelskich właśnie w tych sprawach przed izbą kontroli nadzwyczajnej? Reforma działa i będzie udoskonalana. Dlatego zakres działania Izby Dyscyplinarnej i izby kontroli nadzwyczajnej powinien być rozszerzony. Efekty są widoczne gołym okiem. Do pani Jourovej mam również jedno pytanie. Pani komisarz, gdzie pani była w sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z tego typu nieprawidłowościami.

Mam taką prośbę. Może porównamy system polski do systemu czeskiego. W systemie czeskim sędziów powołuje bez rady sądownictwa prezydent na wniosek ministra sprawiedliwości za zgodą rządu. Sędziowie są powoływani bez udziału rady sądownictwa. To nie sędziowie opiniują sędziów, tak jak to ma miejsce w Polsce. Podkreślam: nie ma rady sądownictwa. Udział rządu, udział prezydenta zamyka całą sprawę. To może w takim razie poprosimy panią komisarz Jourovą o to, żeby udzieliła nam wskazówek, jak zmienić nasz system w kierunku właśnie systemu czeskiego. Jak to jest w systemie czeskim? Minister sprawiedliwości wszczyna postępowania dyscyplinarne bez udziału sędziów. W naszym systemie to wciąż sędziowie oskarżają sędziów, wciąż sędziowie sądzą sędziów przecież. Szanowni państwo, tyle o tym się mówiło, natomiast chciałbym wyraźnie zaznaczyć. Decyzje prezydenta w sprawach powołania sędziów nie mogą być przedmiotem kontroli sądowej. Dlaczego okłamujecie Polaków? Dlaczego chcecie, żeby nasi obywatele byli obywatelami drugiej kategorii w Unii Europejskiej?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia szanuje tożsamość narodową jej państw członkowskich. Skąd to jest cytat? Z naszej ustawy? Nie, to jest tekst wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Radzę się z nimi zapoznać. Dlaczego o tym nie mówicie Polakom?

Dlaczego zakłamujecie rzeczywistość i skazujecie naszych rodaków na podrzędność wobec Niemców, Czechów czy innych Europejczyków? Pozwólcie państwo, że posłużę się drugim cytatem: W myśl art. 4 ust. 2 traktatu Unia szanuje tożsamość narodową jej państw członkowskich, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi. Na temat tożsamości konstytucyjnej i suwerenności wypowiadały się już sądy konstytucyjne wielu krajów, w tym również Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Sprawiedliwości odwołuje się w swoim orzecznictwie do konieczności szanowania tożsamości konstytucyjnej i tożsamości narodowej poszczególnych krajów członkowskich. Kto to powiedział? Dlaczego nie słuchacie swojego eksperta? Co więcej, trybunał ukonstytuował się wówczas jako sąd ostatniego słowa w sprawach ewentualnych sporów z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podkreślam: Brano pod uwagę powyższe, czyli że taki konflikt może nastąpić, więc Trybunał Konstytucyjny zobowiązał się do takiego pojmowania swojej pozycji, że w sprawach zasadniczych o wymiarze ustrojowym zachowa pozycję sądu ostatniego słowa w odniesieniu do polskiej konstytucji. Co takiego stało się przez te lata, że dziś pan profesor zmienił zdanie, a wy prezentujecie stanowisko zupełnie odwrotne? Nie szanujecie konstytucji. Bardzo proszę o szanowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, szanowanie konstytucji i niewprowadzanie naszych rodaków w błąd co do tych kwestii.

Reforma będzie kontynuowana, bo nasi rodacy tego od nas oczekują i dali nam mandat demokratyczny do tego, żeby tę reformę przeprowadzić. Sądy muszą być sprawiedliwe i sprawne. W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej jest znacznie więcej sędziów niż w naszym kraju: we Francji - o 30%, w Hiszpanii - o połowę, w Anglii i Walii - przeszło pięciokrotnie.

Jesteśmy w czołówce krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wydatki. Zarobki początkującego sędziego w naszym kraju to 2,1 średniej krajowej, podczas gdy w Niemczech - 0,9, we Francji - 1,1, w Szwecji - 1,3.

Można by z powodu takich wydatków oczekiwać wspaniałej efektywności ze strony naszych sądów. Tutaj informacja jest nieco bardziej pesymistyczna i negatywna.

Wysoki Sejmie! Dużo w ostatnich dniach było straszenia Polaków tym, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości i następnie wydany wyrok Sądu Najwyższego mogą skutkować unieważnieniem istotnych dla Polaków orzeczeń.

Jednak takie straszenie nie jest pierwszyzną w przypadku totalnej opozycji, bo niestety ta totalność jest wam cały czas bliska.

Takie kłamstwa rozsiewaliście w Europie i musieliśmy konsekwentnie te wszystkie kłamstwa prostować. W związku z jednym z takich kłamstw sąd z Irlandii skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości, czy Polska jest na tyle państwem gwarantującym zasadę niezależności sądów, niezawisłości sędziowskiej, że może wykonywać europejskie nakazy aresztowania. Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział, że sąd państwa unijnego może sprawdzić, czy są gwarancje dla osób poszukiwanych do uczciwego procesu. Straszyliście, że groźni przestępcy nie będą do Polski ściągani na wnioski wynikające z europejskiego nakazu aresztowania.

Zero.

W kilkunastu sprawach ledwie sądy europejskie powzięły wątpliwość, że w Polsce jest jakiś problem z sądownictwem. Wskutek informacji pozyskanych od polskich sądów te wątpliwości zostały rozwiane i poszukiwani zostali wydani. Ba, również w słynnej sprawie irlandzkiej. Straszyliście. Nikt się na te strachy na szczęście nie nabrał, bo żadnego zagrożenia nie było.

Niepokojące z drugiej strony jest to, że przenieśliście skalę swojej narracji, bo przez ostatnie 4 lata mówiliście: konstytucja, konstytucja, zarzucając nam, że ją rzekomo łamiemy. Jednocześnie, kiedy przychodzi do dyskusji o kluczowych prerogatywach wskazanych bezpośrednio w konstytucji, które to prerogatywy nie podlegają kontroli sądowej, jaką jest prerogatywa prezydenta do powołania na urząd sędziego, to już konstytucja przeszkadza. Już prawo unijne jest wyżej, już wyimaginowane kompetencje, których organy Unii Europejskiej nie uzyskały wskutek traktatów, są dla was wyrocznią. Przypomnę państwu szereg orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiadał się o relacji prawa polskiego, konstytucyjnego, z unijnym.

Konstytucja pozostaje zatem - w relacji do traktatu unijnego, akcesyjnego - z racji swojej szczególnej mocy, prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Konstytucja jest najwyżej. Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 konstytucji nadrzędności mocy prawnej korzysta ona na terytorium Rzeczypospolitej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania. Zatem żaden przepis traktatu unijnego, jakkolwiek chcielibyście, żeby rozstrzygał komisarz unijny czy Trybunał, nie może derogować prerogatywy prezydenta. Sprawa relacji polskiego porządku unijnego do krajowego, konstytucyjnego wróciła przy ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Stwierdził w wyroku z dnia 24 listopada 2010 r., powołując się na orzecznictwo niemieckiego trybunału konstytucyjnego, również dotyczące traktatu lizbońskiego, że trybunał niemiecki wskazał, że państwo członkowskie może stwierdzić niezgodność z własną konstytucją aktu prawa unijnego, zachowując prawo do ostatniego słowa. Bardzo jasna jest ta wykładnia. W każdej sprawie, która dotyka porządku konstytucyjnego, to suwerenność państwa i wewnętrzna organizacja konstytucyjna decydują o tym, jak interpretować relacje z Unią Europejską. Polski Trybunał zauważył ten pogląd wyrażany w wyrokach wielu trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich przy rozstrzyganiu tej relacji kompetencyjnej.

Trybunał Konstytucyjny zajmuje się już nie traktatami, ale prawem wtórnym Unii Europejskiej. Nie tym prawem, które wynika z umowy, tylko już stworzonym w Parlamencie Europejskim, w Radzie, w Komisji.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że także ze względu na treść art. 8 ust.1 konstytucji Trybunał Konstytucyjny jest zobowiązany do takiego pojmowania swojej pozycji, że w sprawach zasadniczych, o wymiarze ustrojowym, zachowa pozycję sądu ostatniego słowa w odniesieniu do polskiej konstytucji. Jasno wynika z tego orzecznictwa, że wszelki zbieg kompetencyjny bądź w postrzeganiu kompetencji między państwem członkowskim, w tym przypadku Polską, a Unią Europejską leży ostatecznie w Trybunale Konstytucyjnym. To jest konstytucja, szanowni państwo. Co jest istotne. Pana przewodniczącego Schetyny nie widzę na sali. Nie powtórzy błędów kolegów z wczoraj. Jednak w tym postępowaniu, z którego wyrok zacytowałem, stanowisko zajmował marszałek Sejmu i ówcześnie był nim pan Grzegorz Schetyna. Można przeczytać, że według Sejmu kontrola Trybunału Konstytucyjnego aktów unijnego prawa pochodnego w sprawach wszczętych w drodze skargi konstytucyjnej jest dopuszczalna. Przypominam, że prawo pochodne Unii Europejskiej jest niżej niż traktaty, a w sprawie, o której rozmawiamy, państwo powołujecie się bezpośrednio na traktaty, czyli trybunał jeszcze niższe prawo unijne może badać. Zaczęła się sprawa waszych skarg o polskie sądy do Unii Europejskiej. Ale w międzyczasie również my mówimy: hola, hola. W Niemczech politycy wybierają sędziów. I sąd w Wiesbaden zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Wysoki Trybunale, mnie na urząd powołał minister sprawiedliwości. Ja nie wiem, czy w związku z tym jestem niezawisły, skoro powołał mnie polityk. Ta sprawa znajduje się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jeszcze jest, o dziwo, nierozpatrzona. Trybunał nie zgodził się na połączenie tej sprawy ze sprawą polską. Jednak Trybunał Konstytucyjny Niemiec w jednej ze spraw, która dotyczyła relacji między Niemcami a Unią Europejską, wypowiedział się o relacjach z Unią w zakresie organizacji sądownictwa w ten sposób: Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości przekroczyłby zakreśloną granicę działania trybunału. Jednakże konieczna swoboda w przypisywaniu zadań zawartych w art. 19 ust. 1 akapit 2 traktatu kończy się, gdy interpretacja traktatów nie jest już zrozumiała, a zatem jest obiektywnie arbitralna. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości przekroczyłby tak zakreśloną granicę, działanie trybunału byłoby objęte już art. 19 ust. 1 akapit 2, a orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dotyczące Niemiec nie zawierałoby minimalnego poziomu legitymacji demokratycznej. Czy ktoś krzyczy gerexit? Nie. Wiecie państwo dlaczego? Ponieważ Niemcy szanują swoją suwerenność. Dlatego Niemcy wiedzą, gdzie przekazali swoje kompetencje Unii, a gdzie jest ta granica. A według państwa cokolwiek przyjdzie z Brukseli, jest krytyczne wobec rządu, wobec większości parlamentarnej, to świętość jak Biblia. To jest orzecznictwo wydawane przez wasze autorytety prawne, przez osoby, z którymi chadzaliście tutaj niedaleko z siedziby partii Platformy Obywatelskiej. To jest myślenie niestety prowincjonalne.

Chciałbym w ostatnim słowie odnieść się do. Dziękuję za obecność pana rzecznika praw obywatelskich i możliwość podjęcia dyskusji w ważnych sprawach dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ pan rzecznik poruszył bardzo istotną kwestię. Oczywiście. Poruszył kwestię apolityczności sędziów. Wskazał, że w sprawach polityki rządu czy również ważnych spraw społecznych sędziowie bądź nie powinni się wypowiadać, bądź powinni zachować daleko idącą wstrzemięźliwość. Jak w takim razie skomentować stanowisko stowarzyszenia sędziów Iustitia, które wspierało protest nauczycieli, wydawało stanowiska, odezwy. Przecież, o ile mi wiadomo, protest nauczycieli nie dotyczył prawa do sądu nauczycieli, ale kwestii wynagrodzeń, czyli kwestii kompletnie niezwiązanej z wymiarem sprawiedliwości.

Druga sprawa, ostatnia kampania wyborcza. Tutaj również stowarzyszenie sędziów Iustitia dziwnym trafem, przypadkowo, tydzień przed głosowaniem umieściło serię spotów w Internecie w ramach kampanii straszącej rzekomym łamaniem wolności sądów. Po wyborach już nowych spotów nie było, przed wyborami akurat no zgrało się tak pięknie z kalendarzem wyborczym. Śmiem twierdzić, że przypadkowo, tak jak konferencje prasowe. Rano Platforma Obywatelska zapowiada projekt ustawy o KRS, a w południe przed Ministerstwem Sprawiedliwości sędziowie taki sam projekt proponują. I jeszcze istotna kwestia postępowań dyscyplinarnych i reagowania rzecznika praw obywatelskich na potencjalne naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej. Pan rzecznik bardzo stanowczo zareagował w sprawie pana sędziego Juszczyszyna, który wiemy, że w sposób bezprecedensowy uzurpował sobie kompetencje, których żaden sędzia sądów powszechnych nie posiada. Ale pan rzecznik skorzystał ze swoich uprawnień, podjął reakcję. Dlatego chciałbym zadać pytanie.

Zapytał: Co się stało w Sądzie Najwyższym? Otóż pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani prof. Małgorzata Gersdorf zarządziła wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które się obecnie toczy.

Bardzo dziękuję i oczywiście popieramy ten projekt ustawy.

W dyskusji zgłoszono wniosek o przejście do trzeciego czytania bez odsyłania projektu ustawy do komisji, po doręczeniu posłom zestawienia zgłoszonych poprawek. Do głosowania przejdziemy w bloku głosowań. Wysoka Izbo! Można by było te dwa wystąpienia pana ministra Warchoła i pana ministra Kalety potraktować poważnie, gdyby nie to, że pan marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki upublicznił pismo do marszałka Sejmu, do pani Elżbiety Witek, które skierowała. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Panie pośle, wniosek formalny pan obiecał złożyć. W związku z pismem wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej do pani marszałek Elżbiety Witek, w którym pani wiceprzewodnicząca Komisji nalega na skierowanie projektu do konsultacji do Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy, wnioskuję o przerwę i przygotowanie i skierowanie wniosku Wysokiej Izby do (Dzwonek) Komisji.

Proszę pana posła Tomasza Zimocha o przedstawienie sprawozdania komisji.

Panie Marszałku! Panie Posłanki, Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk. Projekt uchwały złożyli do marszałka Sejmu najpierw Koalicja Obywatelska, następnie klub Lewicy. Obrady były emocjonujące. Jeden z posłów spoza komisji był przeciwny przyjmowaniu takiej uchwały. W czasie obrad pojawiła się propozycja klubu Prawa i Sprawiedliwości, dlatego powołano podkomisję. W czasie jej obrad wypracowany został ostateczny tekst uchwały. W trakcie obrad sprawozdawca wręczył przewodniczącemu w prezencie dwie książki noblistki, by posłowie PiS nie bali się ich lektur, przebrnęli przez nie, zwłaszcza minister kultury i jeden z wicepremierów. Podkreślam bardzo spokojne, kulturalne prowadzenie obrad przez przewodniczącego komisji Piotra Babinetza i podkomisji Jacka Świata. Poseł Ast, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, mógłby naprawdę wiele nauczyć się od swoich klubowych kolegów. Panie pośle, to nie jest pana kompetencja w tej chwili porównywać posłów różnych komisji. Komisja przyjęła treść uchwały przy 25 głosach za i 1 wstrzymującym się. Zatem Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektów uchwał na posiedzeniach w dniach 18 i 19 grudnia wnosi, by Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt uchwały.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji otrzymania przez Olgę Tokarczuk Nagrody Nobla. Polska literatura po raz piąty została wyróżniona Nagrodą Nobla. Do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej dołączyła w 2019 roku Olga Tokarczuk. Autorka 'Biegunów', 'Ksiąg Jakubowych' czy 'Prawieku i innych czasów' odważnie pisze o kryzysie, w jakim znalazła się zachodnia cywilizacja. Mówi, jak trudno dziś scalić świat, który stał się światem fragmentów osobnych, odrębnych bytów i narracji.

Chciwość, brak szacunku do natury, egoizm, brak wyobraźni, niekończące się współzawodnictwo, brak odpowiedzialności sprowadziły świat do statusu przedmiotu, który można ciąć na kawałki, używać i niszczyć. Dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był żywą, nieustannie stawającą się na naszych oczach jednością, a my jego - jednocześnie małą i potężną - częścią' Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie wyrazić uznanie dla Olgi Tokarczuk - laureatki Literackiej Nagrody Nobla za 2018 rok. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża satysfakcję i dumę, że Polska znalazła się wśród ośmiu krajów z największą liczbą Nagród Nobla w dziedzinie literatury.

Bardzo dziękuję, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, bo na razie mamy jedno. Otwieram dyskusję. Jako pierwsza, pani poseł Joanna Lichocka, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Bardzo się cieszę, że udało nam się wypracować kompromisowy tekst uchwały, którą poparły wszystkie ugrupowania oprócz koła Konfederacja. Bardzo się cieszę, że taka okazja jak kolejny Nobel dla polskiej literatury potrafi nas zjednoczyć. To jest duża satysfakcja.

Naprawdę bez względu na to, jak oceniamy poglądy twórców, warto doceniać kunszt, warto docenić warsztat i cieszyć się z tego, że tak prestiżowe nagrody jak Nagroda Nobla przypadają polskiej literaturze. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość oczywiście tę uchwałę poprze. Pan poseł Rafał Grupiński, klub Koalicji Obywatelskiej.

Wysoka Izbo! Radość wielka zawsze, kiedy tego rodzaju zaszczyty nie tyle dotyczą osób, ile dotyczą dzieł, które te osoby tworzą, bo te dzieła w istocie są najważniejsze. Pisarstwo Olgi Tokarczuk to właśnie tego rodzaju wędrówka przez polskie i nie tylko polskie, uniwersalne losy, opisywanie świata w sposób, o którym już tutaj mówiłem, ale o którym warto jedną rzecz powiedzieć, a mianowicie że to jest w jakimś sensie opisywanie czy opowiadanie historii, w której wszyscy możemy się przejrzeć, w której wszyscy możemy się zobaczyć. Kiedyś Józef Korzeniowski powiedział coś takiego, że książki autorzy piszą do połowy, a drugą połowę piszą czytelnicy. Ale wiemy też - państwo po prawej stronie nie lubicie Oświecenia - że Denis Diderot mówił, że kto przestaje czytać książki, przestaje myśleć. Znamy takich, którzy przerwali czytanie, zupełnie niepotrzebnie. Dzięki tej nagrodzie obserwujemy dwa procesy w Rzeczypospolitej. Jeden to wzmożenie, i to jest wzmożenie grafomanów, po prostu ujawniły się setki, jeśli nie tysiące ludzi, którzy nawet potrafili powiedzieć, że Olga Tokarczuk nie jest Polką, że jest antypolska, że jest kimś, za kogo trzeba się wstydzić, wzmożenie pełne, jak mówię, także politycznej grafomanii.

To jest prawdziwy sukces Olgi Tokarczuk, polskiej kultury. Brawo! ...i to jest też oczywiście w jakimś sensie zasługa tych, którzy twórczość Olgi Tokarczuk w akademii noblowskiej dostrzegli.

Dziękuję. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że doszliśmy do konsensusu, i pomimo że ta uchwała nie była procedowana na ostatnim posiedzeniu, tylko jest teraz, cieszę się, że będzie konsensus podczas głosowania. Być może niektórych państwa zdziwię, ale dużo zawdzięczamy tutaj pani Joannie Lichockiej z Prawa i Sprawiedliwości, [[Oklaski]] która akurat czyta książki i rozumie to, o czym mówił wcześniej mój kolega Grupiński i teraz, i na ostatnim posiedzeniu. Tak więc cieszę się, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości podniosą rękę za tym, aby uczcić tę niezwykłą nagrodę Olgi Tokarczuk. Nie chcę wracać do dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu komisji kultury, bo w przypadku niektórych wypowiedzi niektórych posłów była żenująca i nienadająca się do cytowania. Ale z tej mównicy chciałabym powiedzieć, że my, posłanki i posłowie klubu Lewica, jesteśmy dumni całym sercem z tego, że Olga Tokarczuk tak bardzo rozsławiła Polskę na całym świecie. Czytamy jej książki od deski do deski i dla nas było oczywistością to, że Olga Tokarczuk powinna być tutaj w bardzo mocny i bardzo szczególny sposób uznana za perłę polskiej kultury. Chciałabym jeszcze dodać dwa akapity, które nie znalazły się w tej uchwale, a które, uważam, są bardzo szczególne i warto je teraz odczytać. Jako Lewica w swoim tekście uchwały chcieliśmy również, aby zawrzeć takie słowa o Oldze Tokarczuk, że jest to osoba, która uosabia tę część naszej kultury, która nie boi się inności, różnorodności i myślenia poza utartymi schematami, która przekazuje czytelnikowi tę cząstkę prawdy, o której coraz częściej zapominamy, że u podstaw komunikacji między ludźmi leży szacunek i ciekawość, a nie ten sam kolor skóry, wyznanie, te same poglądy czy ta sama orientacja. Ja bym chciała temu posłowi, panu Suskiemu, którego tutaj nie widzę, powiedzieć, że szacunek dla drugiego człowieka nie mierzy się tym, skąd pochodzimy, jaki mamy kolor skóry, co czytamy czy czego nie czytamy. To są podstawowe prawa człowieka, aby szanować każdego. Mówię o tym dlatego, że Olga Tokarczuk szanuje każdego, nawet tego, który nie jest w stanie przeczytać jej książek, i mówi o tym publicznie. Szacunek dla drugiego człowieka jest też czymś, co dla Lewicy jest najważniejsze.

Pan poseł Dobromir Sośnierz, klub Konfederacji. Powiem to, co znaczna część osób na tej sali pewnie myśli w skrytości serca, ale w imię konformizmu boi się albo wstydzi się o tym powiedzieć. Uważam, że recenzowanie różnych wydarzeń przez ciała legislacyjne jest najzupełniej zbędne. Legislatywa jest powołana po to, żeby stanowić prawo, a nie komentować rzeczywistość. Nie ma żadnego powodu, żeby polski parlament opiniował to, czy komitet noblowski dobrze przyznaje nagrody, czy niedobrze. Zwłaszcza w sytuacji kiedy posłowie PiS-u nie znaleźli w sobie odwagi do dzisiaj, żeby podpisać jakże ważne stanowisko odpowiadające Parlamentowi Europejskiemu na jego rezolucję skierowaną do nas, tym bardziej wydaje się niestosowne, żeby wydawać odezwy zupełnie pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Zawsze będę przeciwny temu, żeby Sejm wypowiadał się na tematy pozapolityczne. Gdyby miał taki pomysł, żeby wyrazić uznanie np. dla znakomitych filmów Grzegorza Brauna, to też będę przeciwko. Sejm nie jest od tego, żeby uchwalać, czy Mickiewicz był wielkim poetą albo czy Lech Janerka jest wielkim muzykiem. Zresztą bez urazy, ale rekomendacja tej Izby mogłaby to obrzydzić. Nie widzę powodu, żeby politycy grzali się w blasku cudzych osiągnięć. Próbujecie świecić światłem odbitym, bo sami nie macie, czym się pochwalić. To nie jest żaden patriotyzm, to jest leczenie kompleksów. Jeśli będziemy wypinać się z dumy, że Polak dostał Nagrodę Nobla, to rozumiem, że będziemy też przepraszać, jak Polak kogoś zastrzeli za granicą. Niech każdy wypina własne piersi za własne osiągnięcia i we własne piersi się bije. Założę się, że mniej niż jeden na 100 posłów przeczytał wcześniej jakiekolwiek dzieło pani Olgi Tokarczuk, zanim nie dostała tego Nobla. a nagle czujecie nieodpartą potrzebę wypowiadania się na ten temat.

A państwo chcecie się wypowiadać na takie eleganckie tematy, a tutaj nie potraficie się zachować. Żałuję, że tyle cennego czasu państwo stracili na dopieszczanie tego oświadczenia, w sytuacji gdy nie mamy czasu, żeby się zapoznać z poprawkami dotyczącymi reformy sądownictwa. W dodatku sama twórczość pani Olgi Tokarczuk też budzi moje pewne wątpliwości, więc tym bardziej nie mam powodu, żeby przyłączać się do tych zachwytów. Parę okoliczności świadczy o tym, że tutaj klucz polityczny nie był bez znaczenia przy przyznawaniu tej nagrody.

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Izbo! Przyznanie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk to nie tylko wielkie wyróżnienie i docenienie talentu pisarki, ale też historyczne wydarzenie dla Polski. Jej literatura na wskroś osadzona jest w kontekście polskiej kultury i historii. Jest dziś chyba najlepszą promocją naszego kraju. Mnie osobiście cieszy fakt, że nagrodzona została kobieta wyjątkowa, bezapelacyjnie jedna z najlepszych pisarek, kobieta odważna, która niesie mądre i ważne przesłanie dla współczesnego świata. Jej mowa noblowska powinna trafić do serc każdego i każdej z nas. Jej głos jest próbą zmierzenia się z wyzwaniami, jakie nam stawia teraźniejszość, ograniczaniem praw obywatelskich w imię wyimaginowanych ideologii. Walczy o prawa zwierząt czy wskazuje na konsekwencje zmian klimatu. Takiej wrażliwości i mądrości dziś właśnie trzeba.

Nie będę się grzała w blasku prozaiczki - nie poetki - Olgi Tokarczuk, natomiast mam apel. Na liście lektur jest tylko jedno opowiadanie Olgi Tokarczuk.

Liczę też na to, że w ramach prawie 2 mld zł przyznanych mediom publicznym na rok przyszły zdyskontujemy sukces Olgi Tokarczuk także w mediach publicznych, pokazując ją i na tle pozostałych naszych noblistów, w tym Wisławy Szymborskiej czy Czesława Miłosza, i może także Lecha Wałęsy. Mam nadzieję, że będą to dobre, uczciwe i rzetelne programy publicystyczne i promocja tej twórczości w ramach naszego ogólnonarodowego wstawania z kolan i naszej polityki godnościowej. Wysoka Izbo! Panie marszałku, zwracam się z prośbą o zaproszenie polskiej noblistki Olgi Tokarczuk na najbliższe posiedzenie Sejmu, tak żebyśmy mogli wyrazić ogromne podziękowanie za propagowanie polskiej literatury na całym świecie. Moje pytanie brzmi: Kiedy pan marszałek wystosuje takowe zaproszenie? Dziękuję bardzo. Pan poseł Artur Łącki, klub Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Niestety rzadko nam się zdarza cieszyć z tak wielkich sukcesów naszych obywateli za granicą. I nie dlatego, że są oni mniej zdolni od innych, tylko dlatego, że państwo polskie z twarzą PiS-u nie zorganizowało nic ani nie pomogło nikomu, nie stworzyło żadnych mechanizmów promocji młodych Polek i Polaków w świecie. Za to bardzo dobrze zorganizowało promocję miernych aparatczyków partyjnych w spółkach Skarbu Państwa czy starych aparatczyków partyjnych w fundacji narodowej. Dlatego cieszyć się trzeba z każdego takiego sukcesu na świecie. Pani Joanna Jaśkowiak, klub Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Wyjątkowy dzień, wyjątkowa chwila, krótka - że w takiej zgodzie procedowana jest rzecz, która nas wspólnie, wszystkich, z niewielkim, nieistotnym wyjątkiem, napawa dumą, dumą z Polski, z jej osiągnięć. O ileż przyjemniej byłoby, gdyby wszystko udało się, nawet czasami poświęcając gwałtowność chwili, radość dnia, kiedy żeśmy apelowali o tę uchwałę, na rzecz tej zgody budować. I tak samo byłoby wspaniale, gdybyśmy inne ustawy mogli w tak miłej i zgodnej atmosferze procedować. Tak się niestety nie dzieje. Pozwolę sobie zwrócić się z pytaniem do komisji, czy przewiduje też inne działania upamiętniające tę ważną dla nas wszystkich okazję, czyli Nobla dla pani Olgi Tokarczuk, w tym zaproszenie pani Olgi Tokarczuk do Sejmu. Być może Wysoki Sejm chciałby uczestniczyć w publikacji i promocji dzieł pani Olgi Tokarczuk, jak i innych naszych wybitnych (Dzwonek) noblistów i noblistek. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak pani poseł Nowacka, chciałbym zapytać, czy pan marszałek, pani marszałek przewidujecie zaproszenie do polskiego parlamentu, do Izby niższej naszej noblistki. Warte podkreślenia jest, że w Senacie pan marszałek Grodzki już takie spotkanie odbył. Wydaje się, że również byłaby to idealna okazja do tego, aby pani Olga Tokarczuk mogła wystąpić na tej sali. Dlatego konkretne pytanie: Czy jest taki plan? Czy komisja i pan marszałek planujecie takie rozwiązanie?

Pan poseł Franciszek Sterczewski, klub Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

To jest naprawdę wielki sukces naszej literatury. Wcześniej tu było wspomniane, że to wcale nie jest objaw patriotyzmu, a ja chciałem powiedzieć, że oczywiście jest. To jest wielki sukces polskiej kultury. Olga Tokarczuk jest wspólnym dobrem wszystkich, którzy władają językiem polskim, dlatego to jest nasz wspólny powód do radości. A zatem, szanowni państwo, będąc tutaj, bardzo ciesząc się, że jest sprawa, która może nas połączyć, chciałbym też przyłączyć się do zadających pytanie, czy będziemy mogli (Dzwonek) panią Olgę Tokarczuk gościć w tej Izbie. Pani poseł Katarzyna Kretkowska, klub Lewicy. Wysoka Izbo! Chciałabym zapytać ministra edukacji narodowej, czy rozważa rekomendowanie włączenia większej ilości dzieł Olgi Tokarczuk do lektur szkolnych, bo w tej chwili tylko jedno opowiadanie Olgi Tokarczuk znajduje się na liście lektur w liceach ogólnokształcących. Chciałam też zapytać ministra edukacji narodowej, ministra kultury, może pana premiera o to, czy znajdą się środki w przyszłorocznym budżecie państwa na to, ażeby uzupełnić publiczne księgozbiory, publiczne biblioteki o dzieła Olgi Tokarczuk, gdyż tych dzieł brakuje i w tej chwili Polki i Polacy zapisują się na listach oczekujących, żeby móc te książki w bibliotekach publicznych czytać. Po takim wydarzeniu, wydaje się, państwo powinno wyjść naprzeciw niedofinansowanym bibliotekom publicznym i te książki (Dzwonek) do bibliotek dostarczyć. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke, koło Konfederacji. Panie Marszałku!

Na miejscu tych pól wyrosła dżungla, ta dżungla pochłonęła dwutlenek węgla z powietrza i nastąpiło globalne oziębienie. Oczywiście plotąc takie bzdury, pani Tokarczuk ośmiesza nie Polskę, tylko siebie, ale artyści mogą sobie mówić, co chcą.

Natomiast chcę przypomnieć, że gdyby Sienkiewicz dostawał nagrodę Nobla, to wy byście. wyli z oburzenia, a prawica byłaby tutaj zachwycona, bo on powiedział, cytuję: Prawicę od lewicy dzieli wszystko, również stosunek do znaków arytmetycznych. Prawica uwielbia dodawać i mnożyć, a lewica uwielbia odejmować i dzielić po równo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zamykam dyskusję. Pan sprawozdawca komisji? Do głosowania nad projektem uchwały przystąpimy w bloku głosowań.

Wznawiam obrady. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 104, 105 i 106. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 i 5a regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu przedłożyło projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, druk nr 109. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 102. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawiła opinię dotyczącą wniosku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, druk nr 88. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej sprawy. Kluby przedłożyły wnioski w sprawie wskazania członków Państwowej Komisji Wyborczej, druk nr 92. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej sprawy. Proponuję, aby Sejm podjął decyzję o skróceniu terminu określonego w art. 30 ust. 4 regulaminu Sejmu oraz o rozpatrzeniu wniosków bez przesyłania do właściwej komisji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciw. Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na skrócenie terminu określonego w art. 30 ust. 4 regulaminu Sejm, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Sejm propozycję przyjął. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem wobec rozpatrzenia wniosków bez odsyłania do komisji sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na rozpatrzenie wniosków bez odsyłania do komisji, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Sejm propozycję przyjął. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej, druk nr 108. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 28. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 90. Proszę bardzo. Szczęść Boże! Pytanie brzmi: Czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest krytykiem literatury? Czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest gremium, którego celem jest recenzowanie mądrych bądź głupich werdyktów jakichkolwiek gremiów urzędujących, chwała Bogu, poza granicami Rzeczypospolitej? Państwo nazywacie w swojej uchwale panią Olgę Tokarczuk odważną. Ja nazwę ją koniunkturalistką płynącą na fali poprawności politycznej. Nie żądam uznania mojego punktu widzenia, ale wy, szanowni państwo, nie gwałćcie tej znacznej jednak części narodu polskiego, który rozpoznał w Oldze Tokarczuk kosmopolityczną, antypolską agitatorkę. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie do sprawozdawcy komisji, pani marszałek, i bardzo proszę o to, żeby pan sprawozdawca był uprzejmy odpowiedzieć na to pytanie, o treść tej ważnej uchwały.

Proszę pana posła Tomasza Zimocha o zabranie głosu. Proszę bardzo. Panie pośle, w tej chwili udzieliłam. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panowie Posłowie! Panie Grzegorzu!

O Jezu... „Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji otrzymania przez Olgę Tokarczuk Nagrody Nobla. Polska literatura po raz piąty została wyróżniona Nagrodą Nobla. Do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej dołączyła w 2019 roku Olga Tokarczuk. Autorka 'Biegunów', 'Ksiąg Jakubowych' czy 'Prawieku i innych czasów' odważnie pisze o kryzysie, w jakim znalazła się zachodnia cywilizacja. Mówi, jak trudno dziś scalić świat, który stał się światem fragmentów osobnych, odrębnych bytów i narracji.

Już? Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 90, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 406 było za, przeciw - 1, 17 się wstrzymało. Sejm podjął uchwałę z okazji otrzymania przez Olgę Tokarczuk Nagrody Nobla. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej (druki nr 101 i 108) Proszę pana posła Tomasza Zielińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej. Komisja na posiedzeniu w dniu 20 grudnia, czyli dzisiaj, po przeprowadzeniu pierwszego czytania - tylko dodam, że podczas posiedzenia komisji powstały różne propozycje, czy mamy używać słowa „wysiedleń”, czy „wypędzeń” - i na zasadzie konsensusu uznano, że oba sformułowania znalazły się w proponowanej uchwale. Ostatecznie wszyscy członkowie komisji przyjęli projekt tej uchwały i wnosimy, aby Sejm raczył podjąć tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Panie pośle, czy mogę prosić o odczytanie tej uchwały? Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej. Wybuch II wojny światowej był szczególnie tragicznym doświadczeniem dla ludności Wielkopolski, Pomorza i Śląska oraz innych terenów wcielonych przez Niemców bezpośrednio do III Rzeszy. Eksterminacja elit, masowe wypędzenia ludności polskiej, zasiedlenie tych terytoriów przez Niemców, niszczenie wytworów polskiej kultury oraz grabież polskiej własności związane były z planami całkowitej germanizacji tych obszarów. Te wydarzenia stanowiły realizację nazistowskiej doktryny politycznej zwanej Lebensraum, czyli poszerzenia przestrzeni życiowej narodu niemieckiego. Na Pomorzu niemieckie władze okupacyjne na przełomie października i listopada 1939 r. wypędziły kilkadziesiąt tysięcy polskich mieszkańców Gdyni. Była to pierwsza tak wielka akcja wysiedleńcza przeprowadzona przez Niemców w czasie II wojny światowej. Dla namiestnika utworzonego na terenie okupowanej Wielkopolski przez Niemcy Kraju Warty, Polacy byli: 'elementem niegodnym do włączenia w społeczeństwo niemieckie' Za jeden z początków zorganizowanej, masowej wywózki Polaków uznaje się utworzenie 5 listopada 1939 r. obozu przesiedleńczego na Głównej w Poznaniu, przez który przeszło ponad 33 tys. osób. W pierwszej kolejności wysiedlano ziemian, przedsiębiorców, inteligencję, działaczy niepodległościowych oraz osoby krytykujące niemiecki system nazistowski. Z terenów anektowanych przez Niemcy wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa łącznie niemal pół miliona Polaków, w tym także obywateli Polski pochodzenia żydowskiego i romskiego. Masowe wypędzenia Polaków z terenów Wielkopolski, Pomorza i Śląska oraz innych terenów wcielonych do Rzeszy pozostają bolesnym i wciąż żywym wspomnieniem oraz przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń. W 80. rocznicę pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim ofiarom”

Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Sejm podjął przez aklamację uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 94 i 104) Proszę pana posła Tadeusza Cymańskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Informacja i sprawozdanie są bardzo skromne. Senat przedstawił do zaopiniowania Komisji Finansów Publicznych cztery poprawki. Dwie pierwsze zostały zaopiniowane negatywnie, a dwie następne pozytywnie. Komisja Finansów Publicznych rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tych propozycji i zaakceptowanie ich. Dziękuję bardzo. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywanych poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Poprawki od 1. do 3. zostały zgłoszone do art. 1 ustawy nowelizującej, zawierającego zmianę do ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Do pytania zgłosiła się pani poseł Paulina Hennig-Kloska. Bardzo proszę, pani poseł.

Panie i Panowie Posłowie!

Czy wydaliście więcej, niż mogliście wydać? Ale przede wszystkim chcielibyśmy w końcu dostać odpowiedź na podstawowe pytanie:

Dziękuję, pani poseł.

Wysoka Izbo! Fundusz solidarnościowy miał być takim gwarantem poczucia bezpieczeństwa dla osób, które tutaj, w Sejmie, protestowały, które tutaj, spotykając posłów, pokazywały, jaki jest los dziesiątek tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Przygotowanie tego projektu ustawy przebiegało w sposób haniebny. Te poprawki, które zostały zgłoszone, miały cywilizować projekt. Jesteście państwo przeświadczeni, że nic nie zabieracie. Otóż zabieracie osobom niepełnosprawnym poczucie sprawiedliwości społecznej. Zabieracie poczucie, że osoby niepełnosprawne mogą zawsze liczyć na polski Sejm. I zadaję pytanie: Czy zdajecie sobie państwo sprawę - i pytam pana ministra o to - że te wszystkie osoby w przyszłości będą mogły czuć się oszukane przez polski Sejm, że pieniądze, które miały służyć zapewnieniu im normalności, zostały przekazane na inne cele? Dziękuję, panie pośle. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Proszę o zadanie pytania pana posła Stanisława Pie. Sławomira Piechotę. Przepraszam, to nie mój błąd. Wysoki Sejmie! Kiedy przed rokiem wprowadzano Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, uzasadnieniem dla wprowadzenia nowego podatku oraz przejęcia pieniędzy z Funduszu Pracy była potrzeba wspierania osób niepełnosprawnych. Ta ustawa z nazwy funduszu wykreśla wsparcie osób niepełnosprawnych. I to budzi oczywisty niepokój osób niepełnosprawnych, że ten fundusz przestanie służyć osobom niepełnosprawnym. Senat chce zagwarantować, że pieniądze, które gromadzone są w tym funduszu, będą wydawane na cele służące osobom z niepełnosprawnością. Dlaczego w Komisji Finansów Publicznych PiS głosował za odrzuceniem poprawki Senatu? Na co zatem PiS chce przeznaczyć te pieniądze? Czy to będą dodatkowe pieniądze na propagandę telewizji Jacka Kurskiego?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Pamiętacie może państwo, że wtedy kiedy była podwyższana akcyza na rok 2020, chcieliśmy, żeby te środki były przeznaczone na program walki z chorobami nowotworowymi.

Senat, szanowni państwo, zaproponował, żeby środki z daniny solidarnościowej, środki ze składki na Fundusz Pracy trafiły bezpośrednio do osób niepełnosprawnych.

Wysoka Izbo! Przez przeoczenie.

Dziękuję państwu bardzo. Moje pytanie jest już niestety bezprzedmiotowe, natomiast chciałam powiedzieć, że była to poprawka, która została wypracowana razem z osobami, które reprezentowały środowiska niepełnosprawnych.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Dlaczego większość rządząca nie chce zaakceptować proponowanej przez Senat zasady, która zakłada, że pieniądze z daniny solidarnościowej będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz osób z niepełnosprawnościami? Wszak to państwa posłanka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, pani Urszula Rusecka, przedstawiając Wysokiej Izbie projekt noweli, mówiła, i to jest cytat: wprowadzana nowelizacja ustawy nie ogranicza, nie likwiduje, nie różnicuje wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W podobnym tonie o projekcie ustawy wypowiadał się podczas Komisji Finansów Publicznych pan poseł Cymański. Tu kolejny cytat: Powiedziałem wyraźnie, że pieniądze, które się należą, pieniądze dedykowane z litery i idei, wszystkie trafią do niepełnosprawnych. Dlaczego więc boicie się państwo tej Senackiej poprawki? Czy wcześniejsze deklaracje polityków i polityczek Zjednoczonej Prawicy były po prostu zwykłym kłamstwem? Jeżeli naprawdę zależałoby państwu na zabezpieczeniu praw osób z niepełnosprawnościami, to zagłosowalibyście za Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

W związku z tym Sejm, wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów, poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Pani Iwona Hartwich, Koalicja Obywatelska - bardzo proszę o zadanie pytania. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wczoraj jeszcze państwo dzieliliście się opłatkiem, a dziś pozbawiacie osoby z niepełnosprawnościami szansy na odrobinę lepszego życia. Czym miał być Fundusz Solidarnościowy, to ja doskonale wiem. Powstał on wyłącznie w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami - to była wasza odpowiedź na nasz protest.

Przypomnijcie sobie państwo o tym, kiedy będziecie dzielić się opłatkiem w swoich domach. Jestem waszym wyrzutem sumienia.

Bardzo proszę, pani minister. Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Rzeczywiście to rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pokazał, że tworzy szeroką [[Oklaski]] koalicję na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Proszę pani, to są liczby, które pokazują, jak działamy. Proszę posłuchać spokojnie.

My dzisiaj dajemy 44 mld zł. Szanowni państwo, stańmy w prawdzie, tworząc koalicję na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. My służymy i służyć będziemy osobom niepełnosprawnym.

Skoro odpowiada na pytanie minister konstytucyjny, a państwo tak reagujecie. Czyli rozumiem, że nie chcecie państwo usłyszeć odpowiedzi. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt nie był za, 443 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 95 i 105) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Senat przyjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, uchwalonej przez Sejm 21 listopada. Komisja finansów, po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 19 grudnia, wnosi o odrzucenie uchwały Senatu, a tym samym uchwalenie powyższej ustawy. Dziękuję bardzo. Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu odrzucającą ustawę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci uchwały Senatu odrzucającej ustawę, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu. W uchwale Senat proponuje odrzucić ustawę z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Komisja wnosi o odrzucenie tej uchwały. Do pytania zgłosili się posłowie. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo!

Notariusz może to zrobić nieco szybciej, ale to nie zmieni faktu, że stawiacie przedsiębiorców przed strasznie trudnym zadaniem. Czy to jest droga do normalności, którą zapowiadał pan premier w swoim exposé? Z pewnością nie.

Wysoka Izbo! Korzystając z okazji, że jest pan premier Mateusz Morawiecki, chciałem zadać to pytanie, które się przewija i podczas pierwszego czytania, i podczas posiedzeń komisji, na ostatnim posiedzeniu komisji.

Czy na załatanie dziury budżetowej? Czy z tego tytułu będą realizowane jakieś programy zdrowotne, antyalkoholowe? Takiej odpowiedzi nie otrzymaliśmy do dzisiaj. Pan minister na ostatnim posiedzeniu Sejmu mówił, że nie potrzebuje tych pieniędzy. Jest to zadziwiające. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Rzućcie te papierosy, przestańcie pić alkohol. Nie dajcie Prawu i Sprawiedliwości łatać dziury budżetowej z waszych kieszeni. panie pośle, za bardzo dobrą radę. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Paszyka, Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

żeby pan nam powiedział, jak to jest z tym budżetem. Bo jest dobrze, potem jest źle, potem jest znowu dobrze. Sięgacie do kieszeni Polaków. Sięgacie tym projektem ustawy do kieszeni Polaków, chcecie ich złupić. I tu Wysokiej Izbie by wypadało, panie premierze, wytłumaczyć po co. Po co łupicie Polaków?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 25. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druki nr 96 i 106) Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W wyniku prac komisji, później decyzji Senatu, ta poprawka przeszła.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Prosząc Wysoką Izbę o przyjęcie tej poprawki, chciałabym jednocześnie podziękować Senatowi Rzeczypospolitej (Oklaski), bo dzięki Senatowi Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał 1 mld zł więcej na świadczenia medyczne. Jednocześnie minister finansów może mieć gorzką satysfakcję, bardzo bolesną dla Polaków, bo jeśli PiS przegłosuje dzisiaj ustawę represyjną wobec sędziów, to Polska nie dostanie już żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej (Wesołość na sali), a pan minister nie będzie musiał robić tej ekwilibrystyki. Rząd się wyżywi, może propaganda Kurskiego też, ale na inwestycje nie będzie. Dziękuję, pani poseł. Proszę bardzo.

Szanowni Państwo! Chciałam zadać pytanie, ponieważ. Mówimy w tej chwili o ustawie budżetowej, tak?

Proszę bardzo, pan poseł Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Chciałbym zadeklarować, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest gotowy przychylić się do poprawki zaproponowanej przez Senat, zagłosować za. To zresztą nic dziwnego.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 439 posłów. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Powracamy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 93-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Roberta Telusa o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie!

Ta ustawa jest bardzo potrzebna, oczekiwana przez rolników, przez hodowców trzody chlewnej.

Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 93. Komisje przedstawiają również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

Szanowna Izbo! Nie zgadzamy się, żeby myśliwi wysługiwali się Policją, a taki zapis pojawia się w tej ustawie. Zadaniem Policji nie jest niedopuszczanie nas do lasu, bo właśnie ktoś tam prowadzi odstrzał dzików. Policja ma inne, dalece ważniejsze obowiązki. Dziękuję, pani poseł. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Poprawka dotyczy zapisu, w którym zawarto regulacje dotyczące występowania o pomoc do służb mundurowych w ramach walki z ASF. Krokiem w dobrą stroną jest umożliwienie wystąpienia o taką pomoc w ramach tzw. nadzoru biernego oraz w zakresie kontroli przestrzegania przez myśliwych zasad bioasekuracji w czasie odstrzału sanitarnego. Niestety razem z tymi dobrymi zmianami próbuje się przepchnąć groźny zapis o tym, że myśliwi będą mogli prosić służby mundurowe o zabezpieczenie terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich. Chodzi tutaj o każde polowanie, a nie tylko o odstrzał sanitarny.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

Szanowna Izbo! W tym zapisie proponują państwo, by rokiem więzienia lub grzywną karać osoby, których obecność w lesie w trakcie polowania zostaje uznana za utrudnianie go. Uważamy, że jest to znaczące ograniczenie naszych praw.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Komisje wnoszą o odrzucenie poprawki. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Zalecam spokój. Projekt ten nie zwalcza ASF, bo zamiast koncentrować się na przyczynach rozprzestrzeniania choroby, takich jak brak właściwej bioasekuracji, koncentruje się na eksterminacji populacji dzików w Polsce. Ale cóż jeszcze wprowadza ten projekt? Ten projekt m.in. wprowadza karanie osób, które przeszkadzają w polowaniu. To może dotyczyć również rodzin z dziećmi, które znajdują się na terenie własnej działki albo na terenie lasu. Kiedy znajdą się na terenie polowania, ich również może dotyczyć ta kara. Proszę państwa, to nie jest sposób na pozbycie się ASF-u. To przypomina kolejną ustawę represyjną. I takie ekspresowo uchwalamy już na tym posiedzeniu Sejmu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo! W przedstawionej ustawie proponujecie takie formy przeciwdziałania związane z walką z ASF-em, w ramach których chcecie zamykać przejścia dla zwierząt na drogach i grodzić lasy. To ma fatalne skutki dla całego ekosystemu. Zaburzy to korytarze migracyjne zwierząt. Tak naprawdę, żeby ten zapis był skuteczny, wystarczą maty dezynfekcyjne, połączone z progami zwalniającymi oraz ograniczeniem prędkości na drogach. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości i tożsamej 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości i poprawkę odrzucił. Komisje wnoszą o odrzucenie poprawki.

Wysoka Izbo!

Mam pytanie: Jak państwo to mogli wymyślić i dopuścić do takiego punktu, skoro ten zapis godzi nawet w etykę myśliwych, skoro nawet myśliwi nie są w stanie polować z tłumikami? Co więcej, czy zamierzacie doprowadzić do tego, że zwykli spacerowicze, turyści, miłośnicy przyrody, nie wiedząc, nie słysząc, że na danym terenie trwa polowanie, także mogą stać się ofiarami tej cichej egzekucji? Zapraszam do zadania pytania panią poseł Darię Gosek-Popiołek, Lewica. Szanowni Państwo! To złe rozwiązanie. Tłumiki spowodują, że zwierzęta będą się rozbiegać i płoszyć. Rozwiązanie to jest potencjalnie niebezpieczne dla nas, bo skąd będziemy wiedzieć, że w lesie trwa polowanie. Proszę przypomnieć sobie liczne doniesienia prasowe o tym, co dzieje się na polowaniach. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości oraz tożsamej 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości i poprawkę odrzucił. Poprawki 7. i 8. oraz wnioski mniejszości od 5. do 10. zgłoszone zostały do art. 5 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W 5. wniosku mniejszości do art. 45 ust. 1 wnioskodawcy proponują nowe brzmienie pkt 8c. Nad tymi wnioskami głosować będziemy łącznie. Proszę bardzo, pani poseł Daria Gosek-Popiołek, Lewica. Szanowni Państwo! Chcecie, by właściciele terenów nie mogli decydować o tym, czy na należących do nich terenach będą mogły się odbywać polowania. Chcecie do masowego odstrzału angażować Policję, Straż Graniczną, chcecie zamykać lasy na czas polowania przez Policję. Zadbajmy o bioasekurację, skierujmy tam większe środki, wesprzyjmy rolników, inwestujmy w badania nad szczepionkami przeciw ASF-owi.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wnioski mniejszości odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 7. i 8., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 11. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują skreślić art. 7 projektu ustawy nowelizującej. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo.

Jeden orzeł wczoraj nic nie robił, drugi orzeł dzisiaj się pojawił, nic nie robi. Od 6 lat nie potrafi zrobić ustawy o obwodach łowieckich. Proszę państwa, najpierw trzeba zrobić porządne ustawy o obwodach łowieckich, a dopiero brać się za inne przepisy to regulujące. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. W 12. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują zmianę przepisu o wejściu w życie ustawy. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! W ciągu 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości epidemia ASF osiągnęła takie rozmiary, że zarówno pan minister Jurgiel, jak i pan minister Ardanowski mogą poczuć się ojcami chrzestnymi tej choroby w Polsce. To oczywiście wątpliwa okoliczność do złożenia gratulacji, natomiast znamienne jest to, że przez 4 lata żadne podejmowane działanie nie powodowało jakiegoś znaczącego zastopowania rozwoju tej choroby. Co więcej, prawdopodobnie niektóre podejmowane środki wręcz przyczyniały się do wzrostu ilości problemów. I pytanie do pana ministra Ardanowskiego: Kiedy wreszcie skończą państwo udawać walkę z tą chorobą? Ta ustawa też Policji nakazuje rzeczy, do których Policja nie jest powołana, te wszystkie rzeczy nie wiadomo czy są skuteczne.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub Koalicja Obywatelska zgadza się ze stwierdzeniem, które padło w tej sali z ust pana posła sprawozdawcy, cytuję: Ta ustawa nie rozwiąże problemu ASF w Polsce. Po co w takim razie nam taka ustawa, która nie rozwiązuje problemu? W czasie prac w komisji wykazaliśmy maksimum dobrej woli, zgłosiliśmy wiele poprawek, aby tę ustawę uratować. Odrzucono wszystkie nasze poprawki, co nie pozwala nam w tym momencie poprzeć naszymi głosami tej ustawy. Klub Koalicja Obywatelska będzie głosował przeciwko zaproponowanej ustawie w jej brzmieniu. Dziękuję, panie pośle. Głos ma pan poseł Romuald Ajchler, Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Otóż debatujemy nad ustawą, która tak naprawdę niczego nie załatwia. Ona nie załatwia kwestii likwidacji ASF-u nie tylko w Polsce, ale nie załatwia kwestii tegoż ASF-u w całej Europie, bo my jako kraj nie jesteśmy wyjątkiem, ASF-u nie udało się nikomu jeszcze zlikwidować. Podczas debaty kilkakrotnie zwracałem na to uwagę i pytałem pana ministra, który odpowiadał nam na pytania, pięciokrotnie, czy rząd polski przeznacza jakiekolwiek środki. na badania naukowe, dzięki którym można by wyprodukować szczepionkę, która byłaby skutecznym lekiem na całe zło, które jest dzisiaj w Europie. Jest kilka państw, gdzie ASF-u nie ma, ale to nie znaczy, że go za chwilę nie będzie. Dzisiaj problem ASF-u jest w całej Europie. Panie ministrze (Dzwonek), czy współpracujecie z innymi państwami europejskimi, a także światowymi, aby poszukać skutecznego środka, skutecznego leku? W przeciwnym wypadku tylko odwlekamy to w czasie i męczymy niepotrzebnie także dzikie zwierzęta. Dziękuję, panie pośle.

Wysoka Izbo! Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zwalczać ASF, czy dalej będzie prowadził działania pozorowane? Nie uwzględniliście żadnej poprawki zaproponowanej przez Koalicję Polską - PSL - Kukiz15. To ja w tej chwili pytam was: Co będzie droższe dla budżetu - 500 zł za odstrzelonego dzika, 500 zł za znalezione zwłoki martwego dzika, stworzenie kilku siedlisk dzika czy płacenie z budżetu państwa za utylizowane świnie? W ostatnich 16 miesiącach 50 tys. sztuk świń zostało zutylizowanych. Nie wiecie, skąd wziąć pieniądze? To ja wam podpowiem: z dotacji na TVP, bo Polki i Polacy nie chcą już oglądać niekończącego się serialu pt. „ASF”

Wiemy, że przez 4 lata niewiele działo się ze sprawą ASF-u. Wiemy, że to jest duży problem. Wiemy, że ta ustawa nie jest idealna.

Niemcy wystrzelali 800 tys. dzików. I dało się ten problem ograniczyć. A więc my dzisiaj pomożemy przy tej ustawie i będziemy głosować za. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Chcę bardzo serdecznie podziękować posłom, którzy pracowali nad tą ustawą przez wiele godzin, wykazując troskę i odpowiedzialność za polskie

Chcę odpowiedzieć bardzo prosto i krótko. Choroba, która została wykryta w XIX w. w Afryce, stąd jej nazwa, pustoszy w tej chwili świat: Azję, Europę, pojawia się na innych kontynentach. Choroba jest spowodowana przez bardzo skomplikowany wirus, mutujący wirus, na którego nie ma w tej chwili szczepionki, chociaż prace bardzo intensywnie trwają i Polska jest również uczestnikiem międzynarodowych prac nad znalezieniem szczepionki. Ale tak jak informują najlepsze ośrodki naukowe, jeszcze kilka lat minie, zanim znajdziemy skuteczną szczepionkę zapobiegającą rozprzestrzenianiu się tego wirusa. Choroba jest również w Europie, od Skandynawii po Bałkany, również pojawia się w Europie Zachodniej. W Polsce pojawiła się 17 lutego 2014 r. jako pojedyncze ognisko w pobliżu białoruskiej granicy. Ja mówiłem o tym, bo to jest taki temat dyżurny od tych 5 lat, ponad 5 lat. Może należało zastosować inne metody poprzez ogrodzenie tego terenu i depopulacje zwierząt czy wybicie zwierząt na tym terenie. Może to by przyniosło efekty. Pewności nie ma. W każdym razie ta choroba została rozwleczona na części Polski w województwach wschodnich. Ci wszyscy, którzy zwalczają chorobę, mówią, że są dwa podstawowe działania, które muszą wzajemnie się uzupełniać. Pierwsze to jest bioasekuracja, czyli takie uszczelnienie gospodarstw, żeby wirus z zewnątrz nie dostał się do gospodarstwa. Jako przykład podaje się Hiszpanię, gdzie po 30 latach i wydaniu kilkudziesięciu miliardów euro zlikwidowano praktycznie hodowlę trzody chlewnej we wszystkich mniejszych gospodarstwach, pozostawiając ją na wielkich fermach na pustyni, fermach ogrodzonych drutem kolczastym, odizolowanych jak warowne twierdze, gdzie próbuje się ratować przed zawleczeniem choroby ze środowiska. W Polsce mamy bardzo określoną strukturę gospodarstw również zajmujących się hodowlą trzody, często prowadzoną w starszych budynkach, bez możliwości takiego uszczelnienia tych budynków, żeby ta choroba nie dostała się ze środowiska. Więc trzeba spojrzeć na drugi element, który jest mocno podnoszony również przez Unię Europejską, przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności EFSA. Proszę nie posługiwać się danymi z 2014 r., bo chyba minimalna uczciwość wymaga, żeby posługiwać się danymi, które odnoszą się do czasów współczesnych.

W tym roku mamy 48 przypadków gospodarstw, w roku ubiegłym ok. 210, w latach wcześniejszych wiele, wiele więcej przypadków, czyli choroba w gospodarstwach, o które się najbardziej troszczymy, ustępuje. To pokazuje, że działania, które są podejmowane przez rolników, przez służby weterynaryjne, przez firmy, które również docierają do gospodarstw, są skuteczne. Dość powiedzieć, że od prawie 2 miesięcy nie mamy żadnego przypadku w gospodarstwach. Od 2 miesięcy nie mamy żadnego przypadku w gospodarstwach w Polsce. Natomiast ogromnym problemem jest to, że choroba jest przechowywana w środowisku. Ona jest przechowywana wyłącznie w organizmach dzików. I zalecenie Unii Europejskiej, to, które mówi, że depopulacja dzików do poziomu bezpiecznego jest jednym z nielicznych skutecznych działań, by tę chorobę wyeliminować, chcemy realizować. Oczekiwaliśmy - i tu zawód jest bardzo duży - że instytucja, organizacja powołana do regulowania również populacji zwierzyny, jaką jest Polski Związek Łowiecki, że ta instytucja w trosce i w zgodzie z odpowiedzialnością za polskie rolnictwo, za oczekiwania społeczne takiej depopulacji do poziomu bezpiecznego dokona. Niestety pomimo tego, że część myśliwych dość odpowiedzialnie podchodzi i jest tam wielu ludzi również rozumiejących tę sytuację wojny, na której jesteśmy, wojny z chorobą, to jednak wiele kół łowieckich, wielu myśliwych tych działań nie podejmuje. Dlatego państwo, które chce być skuteczne, nie tekturowe, nie wirtualne, nie teoretyczne, nie może dalej tolerować braku odstrzału, który jest jednym z nielicznych elementów wpływających na likwidację tej choroby. Dlatego podejmujemy ustawę, ustawę specjalną, specustawę, która pozwala państwu uruchomić mechanizmy, których wcześniej nie podejmowano.

Również myśliwi, którzy chcą realizować polowania, zwracają uwagę na działania sprzeczne z prawem, na łamanie prawa przez ludzi, którzy przeszkadzają, utrudniają, uniemożliwiają prowadzenie polowań. Państwo nie może dopuścić do łamania prawa. Łamanie prawa zawsze musi spotkać się z karą.

Proszę państwa, ta ustawa jest tym, czego w tej chwili oczekują polscy rolnicy. Jeżeli ktoś ma do tego oczywiście prawo w demokratycznym kraju, jeżeli będzie występował przeciwko tej ustawie, musi wiedzieć, że działa na szkodę polskiego rolnictwa. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 93, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Nie podałem wyników.

Proszę sprawdzić, panie pośle, czy działa. Tutaj pan chce, Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie projektu ustawy dodatkowo do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest, aby Sejm skierował ten projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu przyjął, a wniosek o dodatkowe skierowanie tego projektu ustawy poddam pod głosowanie. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za dodatkowym skierowaniem projektu ustawy zawartego w drukach nr 45 i 45-A do Komisji Kultury i Środków przekazu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 103. Do pytania zapisał się pan poseł Dariusz Wieczorek, Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście to jest projekt ustawy, który, mówiąc krótko, daje pieniądze i dotacje, które nie będą opodatkowane, polskim obywatelom.

Natomiast pytanie moje jest takie: Czy rzeczywiście dzisiaj jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o realizację ustawy o elektromobilności? Bo przecież zakup samochodów to jest ostatni element, potrzebna jest stacja ładowania, potrzebna jest cała infrastruktura w miastach.

Jako Lewica będziemy głosowali za. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 103, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powracamy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. W trakcie drugiego czytania do projektu ustawy zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. Wobec wniosku o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy bez odsyłania go do komisji po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia poprawek zgłoszono sprzeciw. Odrzucenie tej propozycji będzie oznaczało, że Sejm skierował ponownie ten projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Kto z pań i panów posłów jest za niezwłocznym przystąpieniem do trzeciego czytania projektu ustawy bez odsyłania go do komisji po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia poprawek, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął. Zestawienie zgłoszonego wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawek zostało paniom i panom posłom doręczone do druku nr 107. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 107. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Przed chwilą pan marszałek Senatu Tomasz Grodzki opublikował list Komisji Europejskiej, który został przesłany do prezydenta Rzeczypospolitej, do premiera, do marszałek Sejmu i marszałka Senatu. To jest list, w którym obnaża się te wszystkie kłamstwa, którymi państwo karmicie nas przez ostatnie 24 godziny. To jest list, który mówi prawdę o tym, że po raz kolejny przedkładacie projekt ustawy niezgodny z prawem europejskim i niezgodny z elementarnymi standardami państwa prawa. To jest ostatni moment, byście kolejny raz nie skompromitowali Polski za granicą. To jest ostatni moment, byście kolejny raz nie skompromitowali parlamentu za granicą.

Zapadła decyzja o tym, że przystępujemy niezwłocznie do trzeciego czytania.

Proszę państwa, ja jestem marszałkiem polskiego parlamentu. Uchwalamy w polskim parlamencie prawo.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 1. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują inne brzmienie preambuły. Proszę państwa, jeszcze jedno wyjaśnienie.

Dzisiaj wyraziłam zgodę na 10-minutowe wystąpienia w imieniu klubów. Być może dla państwa hańba, dla mnie - regulamin, art. 182 ust. 2. W 1. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują inne brzmienie preambuły. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Szanowni Państwo! A u kogo nie działa? Można sprawdzić, czy działa.

Proszę państwa, wszystko działa, więc proszę nie wprowadzać marszałka w błąd. Proszę państwa, proszę nie wprowadzać marszałka w błąd. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 3. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie tytułowi ustawy. Przyjęcie tego wniosku mniejszości spowoduje bezprzedmiotowość 4. wniosku mniejszości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 4. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie tytułowi ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przyjęcie tego wniosku mniejszości spowoduje bezprzedmiotowość 1. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przepraszam, Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 18. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 19. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 21. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 20. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 23. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 26. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 27. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przyjęcie tego wniosku spowoduje bezprzedmiotowość 2. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 28. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 29. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 33. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 34. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 35. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 36. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 37. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Z poprawką tą łączy się 12. poprawka. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. i 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 40. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem 43. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 44. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 47. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów jest za przyjęciem 48. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przyjęcie tego wniosku mniejszości spowoduje bezprzedmiotowość wniosków mniejszości od 50. do 56. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 50. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 51. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 52. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 54. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 55. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 57. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują skreślić art. 5. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 57. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przyjęcie tego wniosku mniejszości spowoduje bezprzedmiotowość 9. poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 58. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania, Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 61. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania, Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 60. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tego wniosku spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 11. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W 64. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują skreślić art. 7. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 64. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 68. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 70. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 72. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 73. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 75. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 76. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 77. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 78. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 79. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 80. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 107, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Szanowny Panie Marszałku! Miałem nadzieję, że będę ten wniosek formalny składał, kiedy będzie tutaj pani marszałek Witek, która w trakcie głosowań przed przerwą mówiła o honorze Polski, o szanowaniu polskiego prawa w polskim parlamencie.

Szanowni Państwo! Nie idźcie drogą Marka Kuchcińskiego, bo skończycie dokładnie tak samo. W ten sposób w Polsce ważnego prawa uchwalać po prostu nie wolno. I nie wolno wtedy jeszcze powoływać się na polską konstytucję i na honor państwa polskiego, bo to ani z konstytucją, ani z honorem, ani z państwem prawa.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam wielką przyjemność przedstawić życiorys kandydata do Trybunału Konstytucyjnego pana Rafała Wojciechowskiego, doktora habilitowanego nauk prawnych, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.

W maju 1993 r. ukończył studia i od 1 października tegoż roku został pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji macierzystego uniwersytetu.

W 1998 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez tę izbę. W 2002 r. obronił rozprawę doktorską, a w 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych. Jest autorem dwóch monografii, redaktorem dwóch zbiorów tekstów naukowych napisanych przez wielu autorów oraz autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Uczestniczył w charakterze referenta w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Szczególne zainteresowanie naukowe kandydata po uzyskaniu stopnia doktora budziło sądownictwo polubowne. Historii współczesności arbitrażu poświęcił on kilkanaście publikacji. Jest członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Arbitraż i Mediacja” W 2010 r. został wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W 2011 r. minister sprawiedliwości powołał Rafała Wojciechowskiego na stanowisko notariusza we Wrocławiu. Od 2013 r. kandydat jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2014 r. sprawuje funkcję kierownika Pracowni Europejskiej Kultury Prawnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Analizy Prawa.

W jednym z nich kandydat pełnił funkcję przewodniczącego, a w dwóch - wiceprzewodniczącego.

Proszę pana posła Kamila Bortniczuka o przedstawienie opinii komisji.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Głosujemy nad kolejnymi zmianami w Trybunale Konstytucyjnym w dniu szczególnym. Dzisiaj bowiem zamknął się pewien rozdział politycznej grabieży polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale ten proces zaczął się właśnie 4 lata temu tutaj w polskim parlamencie od brutalnego zamachu, którego dokonał PiS na Trybunał Konstytucyjny. To właśnie wtedy posłowie PiS-u, polski rząd na czele z panią premier Beatą Szydło, zakwestionowali prawidłowy wybór trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W ślad za tym poszły haniebne uchwały.

Później polski rząd zablokował publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego i to był początek wielkiego dramatu, który obserwujemy do dzisiaj. Dzisiaj bowiem o Trybunale Konstytucyjnym nie mówi się jako o bastionie praw i swobód obywatelskich, mówi się jako o bastionie Nowogrodzkiej. Dzisiaj nie mówi się o Trybunale jako o instytucji, do której idzie się po sprawiedliwość, dzisiaj się mówi o trybunale jako o instytucji, do której się chodzi na obiady. Z instytucji wymiaru sprawiedliwości zrobiliście państwo instytucję o charakterze towarzyskim. Mam pytanie do kandydata, chociaż żałuję, że go dzisiaj nie ma z nami. Czy chce pan po koleżeńsku orzekać z prokuratorem stanu wojennego? Czy chce pan po koleżeńsku orzekać z panią poseł, która flagę unijną nazywała szmatą. Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Maria Żukowska, klub Lewicy. Panie pośle, dziękuję panu.

Wysoka Izbo!

Czy uważa, że jest to ustawowa definicja małżeństwa? Prof. Wojciechowski odpowiedział twierdząco na to pytanie, chociaż jako żywo nie jest to definicja ustawowa. W sprawie neutralności światopoglądowej państwa, jak również zasady konstytucyjnej, odpowiedział, że uważa, iż polega ona na tym, cytuję, że nie można pytać o to, kto jest jakiej religii czy wyznania.

W sprawie prymatu prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym pan prof. Wojciechowski uważa, że, cytuję: w Polsce dominuje konstytucja.

Natomiast niestety mogliśmy się przekonać, że nie zna się na prawie międzynarodowym. Nie ma wiedzy ani rozeznania w orzecznictwie TSUE.

Pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Kandydatura pana prof. Wojciechowskiego jest w przeciwieństwie do tego, nad czym głosowaliśmy ostatnio, poważną kandydaturą człowieka o uznanym autorytecie prawniczym, niepochodzącego bezpośrednio z partii politycznej, jak funkcjonariusze, którymi są państwo Piotrowicz i Pawłowicz. Oczywiście pewne obawy budzi fakt, że rekomenduje go Porozumienie, bo boję się, że znowu będzie jakieś rzucanie się Reytanem w sprawach zupełnie niesłusznych i niezasługujących na to, panie wicepremierze. Natomiast jeśli chodzi o meritum sprawy, prawda jest taka, że to, co dzisiaj dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego i to, co dzieje się w związku z sądownictwem, w związku z ustawą o sądach, trzeba powtórzyć, jest to suwerenna sprawa Rzeczypospolitej Polskiej. I to, co dzisiaj już mówiłem z tej mównicy: wara Komisji Europejskiej od tego, w jaki sposób Polacy o swoich sprawach rozstrzygają w tym parlamencie. Wara Komisji i Brukseli od tego tematu. To po pierwsze. Po drugie, trzeba jasno powiedzieć i powtórzyć w tym miejscu, że w 2015 r. zastaliście zabagnioną sytuację i w Trybunale, i w sądownictwie, w całym powszechnym sądownictwie, niesprawiedliwość, wyroki zapadające w skandalicznym trybie, wyroki, które są opóźniane, opieszałość.

Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę pana Rafała Wojciechowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Kto z pań i panów posłów jest za wyborem pana Rafała Wojciechowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Rafała Wojciechowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druk nr 92) Zgodnie z art. 157 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks wyborczy Sejm wskazuje siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Przypominam, że kandydatów na członków Państwowej Komisji Wyborczej wskazują kluby parlamentarne lub poselskie, z tym że liczba tych członków musi odzwierciedlać proporcjonalnie reprezentację w Sejmie klubów parlamentarnych lub poselskich, a liczba członków powołanych w skład Państwowej Komisji Wyborczej spośród wskazanych przez jeden klub parlamentarny lub poselski nie może być większa niż trzech. Na podstawie art. 31b ust. 3 regulaminu Sejmu Prezydium Sejmu ustaliło następującą liczbę kandydatów na członków Państwowej Komisji Wyborczej zgłaszanych przez poszczególne kluby: - Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość - trzech kandydatów, - Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni - dwóch kandydatów, - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) - jeden kandydat, - Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 - jeden kandydat. Proszę o zabranie głosu pana posła Przemysława Czarnka w celu przedstawienia kandydatury pana Zbigniewa Cieślaka zgłoszonego przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana Zbigniewa Cieślaka.

Pan Zbigniew Cieślak jest dobrym kandydatem na stanowisko członka Państwowej Komisji Wyborczej.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana Dariusza Lasockiego. Dariusz Lasocki jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, radnym m.st. Warszawy, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nie należy do żadnej partii politycznej.

Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Międzynarodowym Przeglądzie Politycznym”, „Pulsie Biznesu” Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe. tego kandydata wskazują, iż pan Dariusz Lasocki będzie dobrym kandydatem na stanowisko członka Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę o zabranie głosu pana posła Łukasza Schreibera w celu przedstawienia kandydatury pana Arkadiusza Damiana Pikulika, zgłoszonego przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić kandydaturę pana Arkadiusza Damiana Pikulika. Swoją karierę zawodową zaczynał jako prawnik zatrudniony w kancelariach doradztwa prawnego oraz spółkach prawa handlowego. Prowadzi kancelarię adwokacką. W 2007 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, biegłym sądowym, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu. Zwracam Wysokiej Izbie uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło trzech kandydatów: sędziego, radcę prawnego, adwokata, i to też jest wypełnienie tej dobrej reformy prawa wyborczego, trzech kandydatów, czterech przedstawia opozycja, tak że mam nadzieję, że potraficie to państwo docenić. Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Roberta Kropiwnickiego w celu przedstawienia kandydatur panów Ryszarda Balickiego i Konrada Składowskiego, zgłoszonych przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dwóch bardzo dobrych kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej. Ale też trzeba przypomnieć, jeśli chodzi o system, który zmieniliście państwo w tamtej kadencji, że odchodzimy od systemu sędziowskiego, a przechodzimy na system polityczno-urzędniczy. Jest on dużo gorszym systemem i tak jest powszechnie oceniany w całej Europie. Zawsze urzędnicy... nadzór polityczny nad kluczowymi organami wyborczymi zazwyczaj jest dużo słabszy i organizacyjnie gorszy niż wymiar sędziowski, ponieważ sędziowie, gdy obejmują stanowiska. To bardzo proszę o kandydatury, a nie teraz dyskusję, dobrze? Wyrażam poglądy również kandydatów i myślę, że warto, żeby sala wiedziała, że rekomendujemy bardzo dobrych specjalistów, którzy wiedzą, że system sędziowski, czyli. osób, które powinny nadzorować system wyborczy, które nie są osobiście zainteresowane kandydowaniem i nie mają związków z partiami politycznymi ani instytucjami politycznymi takimi jak choćby Sejm, jest dużo sensowniejszy i dużo zdrowszy dla demokracji. M.in. dlatego nam się udało przeprowadzić tyle elekcji w sposób sensowny i nigdy nie było poważnych protestów i skarg co do ustroju wyborczego. bo nadzorowali to sędziowie. wskazujemy profesorów prawa, wskazujemy specjalistów z zakresu prawa wyborczego, osoby, które mają doświadczenie w. Jak pan nie będzie pokrzykiwał, to będzie krócej. Panu się spieszy, a równocześnie pan przedłuża. Prof. dr hab. Ryszard Balicki jest konstytucjonalistą zatrudnionym na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma na swoim koncie ok. 140 publikacji, w tym publikacje z zakresu prawa wyborczego, takie jak „Zmiana zasad tworzenia okręgów wyborczych w wyborach samorządowych w nowelizacji Kodeksu wyborczego z 2018 r. Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej w świetle regulacji 'Kodeksu wyborczego'” i szereg innych. Jest to człowiek, który bardzo dobrze zna się na organizacji systemów wyborczych i na pracy instytucji publicznych.

To bardzo nowoczesna instytucja, którą tworzył prof. Krzysztof Skotnicki przy współpracy z Państwową Komisją Wyborczą i która zajmowała się i zajmuje do dzisiaj monitorowaniem systemów wyborczych i prawa wyborczego. Konrad Składowski jest osobą, która ściśle współpracuje z tym centrum i jest jego ekspertem. Dr hab. Konrad Składowski jest autorem i współautorem licznych prac naukowych i publikacji z zakresu prawa wyborczego, chociażby takich jak „Kodeks wyborczy, komentarz do zmian 2018” Powinniście przeczytać ten komentarz, bo to jest bardzo dobry komentarz, który jest niestety dość krytyczny w stosunku do tego, co zrobiła Wysoka Izba, jak również ograniczania liczby kadencji, jeśli chodzi o wybory na prezydentów, burmistrzów i wójtów, oraz podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego. Szereg publikacji, które wskazują na to, że te dwie osoby bardzo dobrze znają się na prawie wyborczym i dają rekomendację uczciwego sprawowania funkcji członka Państwowej Komisji Wyborczej i też niezależnego nadzoru nad organizacją wyborów. Bo trzeba pamiętać, że Państwowa Komisja Wyborcza organizuje wybory od najniższych szczebli gminnych po wybory parlamentarne i prezydenckie. Źle się stało, że odchodzimy od systemu sędziowskiego, ale jak już, to trzeba wskazywać osoby niezależne, które mają duży dorobek, i takie osoby wskazała Koalicja Obywatelska. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Gawkowskiego w celu przedstawienia kandydatury pana Liwiusza Laski zgłoszonego przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Wysoka Izbo! Chciałbym zgłosić na członka Państwowej Komisji Wyborczej pana dr. Liwiusza Laskę, który urodził się 22 czerwca 1976 r.

Jest również absolwentem uniwersytetu w Kilonii, gdzie ukończył studia prawnicze. W roku 2011 na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 2004 r. jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego.

Dr Liwiusz Laska jest również prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem prowadzącym praktykę w zakresie procesów sądowych w sprawach prawa pracy, prawa zbiorowego prawa pracy i prawa administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prac legislacyjnych. Jest autorem projektów ustaw, opinii prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego. Doktor Liwiusz Laska od 2005 r. wykonuje zawód adwokata. Był wykładowcą m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Finansów, w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zwracam się do Wysokiej Izby i pana marszałka o to, aby pan Liwiusz Laska został pozytywnie zaakceptowany i wybrany na członka Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę o zabranie głosu pana posła Stanisława Tyszkę w celu przedstawienia kandydatury pana Macieja Miłosza zgłoszonego przez klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie kandydaturę pana Macieja Miłosza na członka Państwowej Komisji Wyborczej. Pan mecenas Maciej Miłosz jest aktualnie radcą prawnym, a zarazem niewykonującym zawodu adwokatem. Uprzednio piastował stanowisko sędziego Trybunału Stanu z woli Sejmu Rzeczypospolitej VIII kadencji. Jest bezpartyjny i nigdy nie był członkiem partii politycznej. Urodził się 18 października 1980 r. w Lublinie.

Od 2010 r. po złożeniu egzaminu adwokackiego nieprzerwanie wykonywał swój zawód adwokata, a następnie radcy prawnego w Lublinie, Stalowej Woli i Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz szeroko pojętego obrotu gospodarczego. Był dwukrotnie zastępcą członka Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Lublinie.

W 2003 r. otrzymał stypendium na uniwersytecie w Gandawie zorganizowane przez ministerstwo do spraw Związku Flamandzkiego Królestwa Belgii.

W przeszłości prawnik w Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa w Lublinie. Członek wielu stowarzyszeń i ich władz statutowych. W latach 2010–2013 członek zarządu, następnie przewodniczący komisji rewizyjnej, zaś od 2016 r. wiceprezes Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie. Od wielu lat poświęca się także działalności pro bono. Pan mecenas Maciej Miłosz spełnia wymagania określone w Kodeksie wyborczym, to jest posiada kwalifikacje równorzędne kwalifikacjom uprawniającym do zajmowania stanowiska sędziego, które już uprzednio piastował w Trybunale Stanu. Jestem przekonany, że zarówno wiedza teoretyczna, jak i bogate doświadczenie zawodowe sprawiają, że pan mecenas Maciej Miłosz jest odpowiednią osobą do piastowania funkcji członka Państwowej Komisji Wyborczej. Bardzo proszę Wysoką Izbę o zaakceptowanie tej kandydatury. Dziękuję. Ponieważ mamy zgłoszenia osób, które chcą zabrać głos w tej sprawie, otwieram dyskusję. Jako pierwszy pan poseł Robert Kropiwnicki. Dziękuję. Jako drugi pan poseł Krzysztof Gawkowski. Również rezygnuje. Dziękuję bardzo.

Proponuję, aby Sejm dokonał wskazania członków Państwowej Komisji Wyborczej w głosowaniu łącznym. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do głosowania łącznego w sprawie wskazania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Kto z pań i panów posłów jest za wskazaniem członków Państwowej Komisji Wyborczej, zgodnie z listą kandydatów z druku nr 92, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm bezwzględną większością głosów wskazał członków Państwowej Komisji Wyborczej: pana Ryszarda Balickiego, pana Zbigniewa Cieślaka, pana Liwiusza Laskę, pana Dariusza Lasockiego, pana Macieja Miłosza, pana Arkadiusza Pikulika i pana Konrada Składowskiego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (druk nr 109) Wysoka Izbo! Zgodnie ze statutem Unii Międzyparlamentarnej członkiem tej organizacji może być cały parlament lub grupa narodowa reprezentująca ten parlament. W poprzednich kadencjach Sejm i Senat były reprezentowane w Unii Międzyparlamentarnej przez grupę narodową.

Prezydium Sejmu proponuje, aby w skład Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej wchodzili wszyscy posłowie Sejmu IX kadencji.

Bardzo proszę. Szczęść Boże raz jeszcze. No jak z tym Noblem? Jak z tym Noblem?

To są korzenie tej organizacji. Pan minister Macierewicz ziewa szeroko, ale nie zajrzał na stronę tej organizacji, na której jest cała globalistyczna agenda. Mamy tam uchodźców nachodźców, rzecz jasna, jako oczko w głowie, mamy tam tęczową rewolucję, [[Oklaski]] niedostatek kobiecości w gremiach parlamentarnych. Cała globalistyczna agenda.

Proponuję, aby Sejm niezwłocznie przystąpił do drugiego czytania projektu uchwały. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do drugiego czytania. Pan poseł jeszcze raz. Pół minuty, panie pośle. Kiedy projekt Unii Europejskiej był jeszcze mały, zalążkowy, jeszcze to nie śmierdziało eurokołchozem, jeszcze to nie było totalniackie na tę miarę, jaką osiąga dzisiaj, miarę absurdu oczywiście, wtedy niektórzy myśleli, że to jest jakaś miła międzynarodówka troszkę Żydów, troszkę masonów, troszkę eurokomunistów. Wszyscy myśleli, że to takie niewinne. A oto dzisiaj Lewiatan, szanowni państwo, wyciąga nie wiem jaką tam kończynę czy ogonem macha i zamiata polską suwerenność. Nie wchodźcie w projekty, które z daleka zalatują masońskimi priorytetami pacyfizmu, globalizmu.

Kto z pań i panów posłów jest przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 109, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 102) Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 102, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Ogłaszam 3-minutową przerwę.

Wysoka Izbo! Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że do wygłoszenia oświadczeń poselskich zgłosił się jeden poseł. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenia? Dobrze, czyli dwie osoby. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam za zamkniętą.

Wysoki Sejmie! Dobrze, że dużo mówi się o godnym upamiętnieniu triumfu Polaków nad bolszewikami w 1920 r. Najczęściej wspomina się o łuku triumfalnym, który miałby upamiętniać tamto wydarzenie. Wydaje się jednak, że potrzebny jest nam głębszy namysł, abyśmy nie popełnili błędu, który byłby znakiem braku wdzięczności, a przynajmniej błędem spłaszczenia własnej historii. Bitwa o Warszawę przypomina bardzo bitwę o Wiedeń. Tam Europie zagrażali Turcy, tutaj bolszewicy. Czy tylko? Polski król Jan III Sobieski, pokonawszy Turków, nie przypisał zwycięstwa sobie. Powszechnie znana jest jego parafraza słów Gajusza Juliusza Cezara: Veni, vidi, vici.

Tak skromność króla uratowała w 1683 r. Europę od fanatyzmu islamskiego. Zarzucano królowi, że nie wykorzystał wiktorii wiedeńskiej, aby uczynić Polskę krajem dominującym w Europie. On jednak w swojej mądrości wolał przegrać bitwę dyplomatyczną i zadowolił się zwycięstwem w boju o Wiedeń i cały kontynent. Udało mu się odkryć drogę, którą wyznacza Pan Dziejów. Gorzej jest z nami i cudem nad Wisłą. Od początku nie chciano uznać, że tutaj też stało się coś wyjątkowego. Zwyciężaliśmy kolejny raz, nie siłą oręża, ale ducha. Na ten temat zgromadzono wiele świadectw. Mówili o tym nie tylko żołnierze polscy.

To Matka Boska na niebie widziana była przez setki bolszewików, to jej pojawienie się na niebie w otoczeniu husarii, polskiego zwycięskiego wojska, które pod Wiedniem z hasłem: W imię Maryi rozegnało pogańskie watahy, wywołało wśród sołdatów strach, przerażenie i panikę, której nie sposób opisać. Tak o końcu marszu bolszewików na podbój świata mówili uczestniczy tamtych wydarzeń. Naród wytężył wszystkie siły, nie sposób pominąć zasług marszałka Józefa Piłsudskiego, sztabu generalnego, dowódców, żołnierzy, wszystkich obrońców ojczyzny, ale wtedy cały naród zjednoczył się w potężnej modlitwie, wołając do swojej królowej o ratunek i do Boga o zmiłowanie nad zagrożoną Polską. Czy łuk triumfalny uwzględni te dwa czynniki zwycięstwa: ludzki i ten dominujący - boski? Czy dalej będziemy udawać, że oświeconym Europejczykom nie wypada mówić o cudach? Czy taka degradacja zdarzeń przystoi ludziom wierzącym i praktykującym? A może ktoś z projektantów monumentu zainspiruje się obrazem, który został namalowany na ścianie kaplicy Castel Gandolfo, przedstawiającym cud nad Wisłą?

Widać tam walczących żołnierzy, księdza Skorupkę i interwencję nieba. Może w tym źródle i w tym zwycięstwie trzeba szukać klucza do rozwiązania naszej trudnej sytuacji? Potęga ducha jest zawsze wyżej niż wszelka doczesność. Ognia, który tli się w narodzie, 100 lat nie wyziębi i tylko czy ten ogień, prawda, dobro narodu i ojczyzny jest jeszcze w kręgu naszych marzeń? Dziękuję bardzo. Zapraszam panią poseł Elżbietę Płonkę, Prawo i Sprawiedliwość, do wygłoszenia. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Niedługo Warszawę czekają podwyżki za odbiór odpadów uchwalone przez rządzącą miastem Koalicję Obywatelską. Podwyżki oczywiście zaproponował prezydent Rafał Trzaskowski. Kto jest winien tej sytuacji? Zdaniem prezydenta Trzaskowskiego za skalę podwyżek za odpady, z którymi teraz mierzą się miasta i gminy w całym kraju, odpowiada wyłącznie rząd Prawa i Sprawiedliwości. No to przyjrzyjmy się, jak funkcjonował dotychczasowy system odbioru odpadów komunalnych w Warszawie i jaka jest rzeczywista przyczyna podwyżek. W lipcu 2012 r. weszły w życie przepisy stanowiące, że śmieci i różnego rodzaju odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych stanowią własność gmin. Miasto stołeczne Warszawę podzielono wówczas na 9 rejonów, w których odpady miały odbierać firmy wyłonione w przetargu. Całość operacji wiązała się z wprowadzeniem opłat za wywóz śmieci, które miały być liczone od osoby w budynkach wielolokalowych. Okazało się, że taki system oznacza podwyżkę dla gospodarstw domowych. System ten okazał się nie tylko drogi, ale także niewydolny. Jedna z firm obsługująca trzy z tych rejonów w miesiącach letnich przestała w wyznaczonych terminach odbierać śmieci. Zgodnie z możliwościami, jakie daje prawo, gminy mogą z odpadami komunalnymi zrobić kilka rzeczy. Najbardziej pożądaną sytuacją, do której samorządy powinny dążyć, jest stworzenie systemu instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, potocznie zwanego recyklingiem. Niestety większość odpadów z Warszawy nie trafia do tego systemu. Przez 6 lat m.st. Warszawa, które posiada własną spółkę, MPO, nie stworzyła własnego systemu przetwarzania odpadów komunalnych, takiego jaki np. jest w Krakowie. Inną możliwością, z której mogłaby skorzystać Warszawa, jest budowa nowoczesnej spalarni odpadów. A obecnie istniejąca spalarnia odpadów nie jest w stanie zaspokoić potrzeb miasta. Najmniej pożądaną i jednocześnie najdroższą formą gospodarowania odpadami jest ich składowanie. Warszawa właśnie taką formę gospodarowania odpadami wybrała. Tymczasem jedno z głównych miejsc, dokąd wywożono odpady Warszawy, czyli składowisko odpadów Radiowo w gminie Stare Babice, zostało decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska zamknięte. Decyzję tę podtrzymał także sąd administracyjny. Na to składowisko skarżą się szczególnie mieszkańcy Bemowa, Żoliborza i Bielan, ponieważ w przypadku wiatru zapachy z wysypiska odczuwane są w tych dzielnicach. Co to wszystko oznacza? Od 2012 r. większość śmieci wbrew zaleceniom ląduje na wysypiskach odpadów, a tylko niewielka ich ilość trafia do systemu przetwarzania odpadów komunalnych. W wielu państwach świata gminy zarabiają na przetwarzaniu odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych, ale niestety w europejskiej stolicy, jaką jest Warszawa, prezydent Trzaskowski postanowił sięgnąć do kieszeni warszawiaków, aby pokryć niedobory związane z nieudolnością urzędu, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami. Prezydent Trzaskowski twierdzi, że za wzrost opłat za odbiór odpadów odpowiada min. wzrost opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska. No skoro władze Warszawy, zamiast tworzyć system przetwarzania odpadów komunalnych, zajmowały się tylko upychaniem śmieci po sąsiednich gminach, to nie jest dziwne, że opłata marszałkowska dotknie Warszawę. Można tego uniknąć, ale trzeba przetwarzać odpady, a nie je składować, opłata marszałkowska bowiem wzrasta nie za odbiór odpadów - nie wzrasta za ich przetwarzanie, nie wzrasta za ich spalanie - ona wzrasta właśnie za składowanie. Ponadto co się stało z pieniędzmi, które warszawiacy wpłacają do kasy miasta za wywóz odpadów komunalnych? Przecież przez 6 lat Warszawa z tytułu opłat musiała zebrać kilkaset milionów złotych. Gdzie są te pieniądze? Co się z nimi stało? Czy nie można było za te pieniądze rozpocząć budowy systemu recyklingu? A więc przyczyną podwyżek nie są działania rządu, który musi dostosować gospodarkę odpadami do norm unijnych, ale wieloletnie nieróbstwo, lenistwo i zaniedbania władz Warszawy. Pan prezydent Trzaskowski zamiast skarżyć się na rząd i zamiast podnosić ceny odbioru śmieci, powinien jak najszybciej przedstawić plan stworzenia systemu recyklingu dla Warszawy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę o wygłoszenie oświadczenia. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przyjęliśmy dziś ustawę o ustroju sądów powszechnych w ramach reformowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Chcę zwrócić się do wszystkich wykonujących zawód związany z wymiarem sprawiedliwości - jest to jednak trzecia władza, a przecież jest jeszcze władza ustawodawcza i wykonawcza. Wielu sędziów, jak pokazuje obecny czas, usiłuje postawić władzę trzecią nad pierwszą i drugą konstytucyjną władzą. Ja, jako lekarz medycyny i polityk, nie rozumiem tej wyjątkowej sytuacji wytworzonej przez grupy sędziów tworzących reguły państwa w państwie. Wykonując mój zawód, nie jestem wyłączona z ponoszenia odpowiedzialności w moim postępowaniu za zdrowie i życie ludzkie, nie mogę narzucać swoich poglądów ani decyzji choremu człowiekowi, ponoszę też odpowiedzialność deliktową, o której muszę pamiętać. Jak to jest, że sędzia, prokurator, nie mówiąc o adwokacie, może postępować według własnych reguł wobec spraw ludzkich, które mają wagę nawet większą niż zdrowie? Bywa, że ludzie są krzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, zostają pozbawieni zdrowia i środków do życia wskutek niesprawiedliwych wyroków, a nawet umierają z tego powodu, że zostali takimi wyrokami bardzo skrzywdzeni. Jaka jest odpowiedzialność tych osób za wyroki godzące w sprawiedliwość? Czy pytanie o sumienie sędziego ma tu w ogóle sens? Niestety pozostawienie wymiaru sprawiedliwości bez dekomunizacji i brak przepisów prawa dyscyplinujących sędziów sprawia, że woła się z polskiej ulicy o ratunek, o państwo prawa.

Wyjaśnienia sędziego rozpatruje trzech sędziów, kolegów z tego samego sądu. A stwierdzenie: autorytet moralny sędziego przemawia za wiarygodnością złożonego wyjaśnienia, brzmi jak: samooceniający się autorytet. To rzeczywiście wyjątkowy samoautorytet, niczym w kaście bogów olimpijskich. Kto z ludzi wkraczających na salę sądową po sprawiedliwość może na nią liczyć, jeśli sędzia jest nieomylny, jeśli jest pewien swojej niepodważalnej decyzji? Wielu pokrzywdzonych ludzi w Polsce szuka sprawiedliwości i woła do rządu o ograniczenie samowładzy i hermetyzacji kasty oraz obstrukcji sędziowskiej. Jest to wielka bolączka sądów, a bywa, że idą za tym nieprawidłowe decyzje prokuratury ze względu na zależności personalne. Rząd Zjednoczonej Prawicy ma obowiązek dokonywać zmian ustrojowych w imię demokratycznie udzielonej władzy przez Polaków oczekujących sprawiedliwości może bardziej niż chleba powszedniego. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj na naszym posiedzeniu przyjęliśmy przez aklamację poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej. I bardzo dobrze, bo takie daty powinno się pamiętać i takie rzeczy powinno się czcić i chwalić. Przepraszam, nie chwalić, tylko pamiętać o nich, bo one nas scalają i czynią to, że jesteśmy silniejsi jako naród. Ale ja jako wnuk i syn Sybiraków mam obowiązek z tej trybuny powiedzieć i przypomnieć posłom z Komisji Kultury i Środków Przekazu i wszystkim posłom Rzeczypospolitej, że 10 lutego 1940 r. rozpoczęły się pierwsze wywózki obywateli polskich na Sybir i że już za 2 miesiące będzie 80. rocznica tych pierwszych wywózek. Z tej trybuny proszę zatem posłów o to, abyśmy taką samą uchwałą uczcili pamięć ludzi, którzy zostali wywiezieni na tą nieludzką ziemię, tych, którzy wrócili, jak również tych, szczególnie tych, którzy tam zostali. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska.

Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny 3. posiedzenia Sejmu, zwołanego na dni 8 i 9 stycznia 2020 r., został paniom i panom posłom doręczony.